Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bronisław Cieślak - wielka postać polskiej kultury. Dla wielu Polaków był przede wszystkim lubianym i cenionym aktorem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Grał w jednym z najbardziej znanych polskich seriali. Kultowa rola Sławka Borewicza z serialu „07 zgłoś się” towarzyszyła milionom Polaków i w młodości, i w starości. Był również politykiem. W roku 1997 r. uzyskał mandat poselski z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W III kadencji zasiadał w komisjach administracji i kultury. Klub Lewicy będzie go przede wszystkim pamiętał jako zaangażowanego i sprawnego człowieka kultury, osobę, która dla polskiej kinematografii zrobiła bardzo dużo. Pamiętamy, że był rzecznikiem klubu parlamentarnego.

Bliskim składamy wyrazy współczucia. Prosimy o minutę ciszy.

Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatu pani poseł Anny Wasilewskiej na podstawie art. 251 § 5 Kodeksu wyborczego postanowiłam o wstąpieniu na jej miejsce pani poseł Anny Wojciechowskiej, która zgłosiła się do ślubowania poselskiego. Panie i panów posłów proszę o powstanie. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Pani poseł Anna Wojciechowska. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pani poseł Anna Wojciechowska złożyła ślubowanie poselskie. Obecnie, proszę państwa, przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa obecnych na sali, a także tych, którzy łączą się z nami zdalnie, o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Rozumiem, że sprzeciw wobec tego, że koło ma 5 minut, tak? Dobrze.

Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1131. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Informuję, że w związku z niezgłoszeniem przez uprawnione podmioty tematu informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących punkty te nie zostaną rozpatrzone na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Wczoraj stała się rzecz niesłychana, wczoraj pan minister Buda, który jest odpowiedzialny za Krajowy Plan Odbudowy, wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że Krajowy Plan Odbudowy został wysłany do Brukseli, że już nic nie można zmienić - w przeddzień debaty w parlamencie, w przededniu zakończenia negocjacji przez samorządowców. Dzisiaj trzeba zadać jedno, najważniejsze pytanie: To po co jest parlament? Gdzie jest podmiotowość parlamentu, o której tyle razy mówiliście, do której tyle razy się odnosiliście? Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest wyjątkowa, bo tak naprawdę doszło do wielkiej zdrady polskich samorządów i ludzi, jeżeli chodzi o zakres Krajowego Planu Odbudowy. I wy to zrobiliście razem z PiS-em, droga Lewico.

Wniosek przeciwny, proszę państwa. 2 miesiące trwały konsultacje. Platforma nie była w stanie się zdecydować, jak będzie głosować. Teraz pan przewodniczący wychodzi i opowiada bajki, że nie było możliwości konsultacji. Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Minuta, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Decyzja pana premiera o podpisaniu się pod Funduszem Odbudowy w ubiegłym roku to jedna z najważniejszych decyzji od czasów traktatu lizbońskiego. I zanim przejdziemy do przyjmowania lub odrzucania tego funduszu, do głosowania nad nim, Sejm powinien ustalić, jaką większością będzie przyjmowany Fundusz Odbudowy. Dysponujemy opiniami, które mówią, że ta zmiana wymaga większości 2/3 głosów, [[Oklaski]] ponieważ jest przekazanie kompetencji państwa członkowskiego na rzecz instytucji europejskich w zakresie podatków i wypuszczania wspólnych obligacji, jest przekazanie kompetencji konstytucyjnych ministra finansów.

Art. 90 ust. 1 mówi o przekazaniu uprawnień suwerenności komisji. Nie mamy z tym do czynienia, państwo doskonale o tym wiecie. Dysponujemy sześcioma opiniami prawnymi, nie tylko Biura Analiz Sejmowych, ale także opiniami zewnętrznymi, które wyraźnie mówią o zwykłej większości. W związku z tym nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo musiałabym z premedytacją złamać konstytucję.

W związku z tym nie poddam tego pod głosowanie. Proszę bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym jednak złożyć wniosek, żeby rozpatrzyć, czy wniosek pani marszałek jest słuszny czy niesłuszny. Przy okazji chciałbym zauważyć, że gdyby jakiś poseł czy senator I Rzeczypospolitej wziął od Prusaków czy Rosjan worek złota za coś tam, za jakieś głosowanie, i rozdał ten worek. Mówię to do posłów Lewicy. Proszę bardzo, wniosek formalny - mam nadzieję - pani poseł. Panie pośle, to nie jest wniosek formalny, więc może mi pan to zostawić na wieczną pamiątkę, chętnie się z tym zapoznam. Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek formalny o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad informacji pana premiera o obecnym kształcie Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedzieliśmy się, że to, co zostało wysłane do komisji, jest jakąś roboczą wersją z piątku.

Tak z ludzkiego szacunku i z ludzkiej grzeczności, panie premierze, warto, żeby pan odpowiedział nam na pytania. Dziękuję, pani poseł. Pan premier jest na sali. Będzie za chwileczkę możliwość zabrania głosu przez wszystkie kluby. W związku z tym, że został zgłoszony wniosek formalny o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Państwo Ministrowie!

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska i Koło Poselskie Konfederacja złożyły wniosek o wysłuchanie publiczne. W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony przez połączone komisje. Do projektu ustawy zgłoszono ponadto sześć poprawek. Biuro Legislacyjne wyraziło swoje formalne zastrzeżenia co do zasady poprawek zgłaszanych do ustawy ratyfikacyjnej. Ze względów proceduralnych poprawki zostały poddane pod głosowania. W głosowaniu nad całością rządowego projektu ustawy z druku nr 1130 ustawa uzyskała zdecydowane poparcie posłów. 53 osoby głosowały za ustawą, trzy osoby były przeciwne, a pięć osób wstrzymało się od głosu. Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył przedmiotowy projekt ustawy, ustawy bardzo ważnej dla Polski i Polaków. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 17 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dzisiaj, w przededniu tak ważnej decyzji, trzeba przypomnieć o tym, jak bardzo mocno tamta decyzja oparta była na szerokim konsensusie społecznym.

Podczas tego głosowania, które jest przed nami, będziemy mogli wyrazić się mocno, opowiedzieć za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej, za wykorzystywaniem środków, które będą nam przekazywane do dyspozycji, bądź wyrazić wobec tego sprzeciw.

Ale trzeba też w tym kontekście powiedzieć, że bardzo szybko te cele zostały uznane przez wszystkie kluby parlamentarne, przez wszystkie partie, przez prawie wszystkie partie, przez zdecydowaną większość. To były cele, które nas przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci, można powiedzieć, łączyły. Dziś zatem powiedzmy raz jeszcze głośne „tak” dla rozwoju Polski, głośne „tak” dla rozkwitu Polski, również dzięki środkom unijnym. To duża szansa na szybkie wyjście z pandemii, szybkie wyjście z COVID-19. Zacznę od tego, że dzisiejsza ustawa, którą tutaj przedkładamy, która ma na celu zatwierdzenie możliwości korzystania ze środków unijnych, była negocjowana parę lat, a ostatnie kilkanaście miesięcy to był bardzo burzliwy proces. Otóż najbardziej przeciwni byli zachodni politycy i zachodni ekonomiści, którzy nie chcieli przekazywać środków netto dla Polski, dla krajów Europy Środkowej.

Dlatego z całą mocą, także ze wsparciem krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych państw Europy Środkowej, kładliśmy na to nacisk, mówiąc, że te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych, jeżeli chodzi o wyjście, szybkie wyjście z COVID-19, żeby z powrotem ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju Unii Europejskiej, rozwoju gospodarczego. Potem po tych długich negocjacjach, po zatwierdzeniu w Radzie Europejskiej nastąpił proces konsultacji. O te konsultacje państwo tutaj dopytywaliście.

Były spotkania, w których uczestniczyłem osobiście, również w komisji wspólnej rządu i samorządu. Była także Rada Dialogu Społecznego, były spotkania z przedsiębiorcami, liczne spotkania z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorcami rolnymi. To wszystko były wielodniowe dyskusje dotyczące poszczególnych zapisów Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkim organizacjom pozarządowym, wszystkim województwom, z którymi był ten program konsultowany, szeroko konsultowany, bardzo serdecznie dziękuję za liczne uwagi, za liczne propozycje. Chcę powiedzieć, że wiele, bardzo wiele z nich zostało ujętych w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego dzisiaj warto podkreślić z całą mocą, Wysoka Izbo, że to nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie. To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom - może szpitalom, w których leczy się ktoś bliski z państwa rodziny, może szkołom, w których uczy się któreś z państwa dzieci - które mają pomóc Polakom w otrzymaniu szansy na lepszą infrastrukturę: drogową, kolejową, internetową, energetyczną. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski. I dlatego bardzo gorąco apeluję do wszystkich sił politycznych: odłóżmy swary, kłótnie, odłóżmy tę logikę: oko za oko, ząb za ząb. Dzisiaj apeluję do wszystkich klubów politycznych: przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski, ponieważ ta ustawa, za którą stoją te środki unijne, jest rzeczywiście ustawą o polskiej racji stanu.

Ta ustawa o środkach własnych to ustawa o przyjęciu bądź nie środków unijnych na polski rozwój, na polski rozwój na najbliższą dekadę. Ta decyzja jest jedną z najważniejszych decyzji na najbliższe 10, 20 lat.

nie pozwolili, żeby kryzys gospodarczy dotknął ich tak, jak dotknął inne kraje w Europie, ale sami siebie postanowili skrzywdzić poprzez brak przyjęcia tak wielkich środków netto. Podkreślam: te środki to nie tylko krajowy program odbudowy, to ponad 700 mld zł, w cenach bieżących to ok. 770 mld zł dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy. Nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marshalla. Nie wolno też, szanowni państwo, igrać z taką szansą, bo rzeczywiście ona jest bezprecedensowa.

Dlatego chcę z całą mocą podkreślić: dzisiaj przezwyciężmy te nasze podziały. Bo tutaj nie chodzi o tę czy inną rację polityczną czy rację partii politycznej, chodzi o polską rację stanu. Zagłosujmy za polską racją stanu. Pytaliście państwo o konkretne środki. W procesie konsultacji wszystkie te środki bardzo łatwo jest zdekomponować, podzielić na powiaty, miasta, gminy. Można zadać takie pytanie: Czy właśnie np. mieszkańcy Wielkopolski nie potrzebują 70 mld zł w najbliższych kilku latach na rozwój dróg, infrastruktury i wiele innych celów? Oczywiście potrzebują. Czy mieszkańcy Gdańska nie zasługują na ponad 9 mld zł w kolejnych kilku latach z tych wynegocjowanych przez nas programów? Oczywiście potrzebują ich i zasługują na nie. Albo mieszkańcy Warszawy - ponad 30 mld zł. Albo mieszkańcy powiatu gorlickiego - 2 mld zł przez najbliższych kilka lat. Nie odrzucajcie tych środków dla mieszkańców naszych powiatów i gmin. To wielkie dzieło nie może być przedmiotem hazardu, nie może być przedmiotem różnych sztuczek, kuglowania czy partykularyzmów politycznych, bo będzie to przypominać rosyjską ruletkę. Z tym że pistolet wymierzony jest wtedy w Polaków, w polskich przedsiębiorców. Nie można igrać w ten sposób z wielką szansą rozwojową, przed którą stoimy. Drodzy Państwo!

Wtedy duża większość ówczesnych parlamentów przegłosowywała te środki, wiedząc, że jest to znakomita szansa rozwojowa, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma tutaj do czynienia z igraniem, z ryzykowaniem tymi wielkimi szansami rozwojowymi, w tym dla Polski.

A więc mówimy o rzędzie wielkości daleko mniejszym. To ponad rząd wielkości mniej niż to, co wcześniej było uważane za środki unijne. Ale powiedzmy sobie też dodatkowo, jak one mają być spłacone, bo tutaj też niektórzy starają się siać ferment i wprowadzać w błąd. Otóż nie ma tu, szanowni państwo, żadnego uwspólnotowienia długów. To znowu argument ekonomistów niemieckich, holenderskich, belgijskich, austriackich i duńskich. Oni nie chcą tego funduszu, bo oni muszą netto do niego dokładać. Dlatego nie ma tu uwspólnotowienia. Jest mechanizm grantowy oraz mechanizm pożyczkowy, jeżeli z niego skorzystamy.

Czy zatem nie warto jest skorzystać z wielkich środków teraz, kiedy gospodarka globalna została tak fundamentalnie poszkodowana poprzez COVID-19, żeby wyjść z tego kryzysu jak najszybciej? Nie ma ryzyka ciążącego na Polsce, że będziemy spłacać długi Włoch czy Francji. Szanowni państwo, chciałbym, żeby Polska była jak najszybciej na poziomie rozwoju Francji czy Włoch. Właśnie te środki do tego służą. Służą one do tego, żebyśmy jak najszybciej, jak najlepiej mogli rozwinąć naszą gospodarkę i żebyśmy mogli doścignąć tych najlepszych. Dlatego w tym procesie konsultacji, dyskusji chciałbym też podziękować. Chciałem podziękować wszystkim, którzy skierowali swoje merytoryczne uwagi. Chciałem podziękować klubowi Lewicy, bo przekazał nam najbardziej kompleksowy dokument, długi, 80-stronicowy merytoryczny dokument. Chcę powiedzieć, że ten rzeczowy, merytoryczny dialog z Lewicą zaowocował włączeniem do programu odbudowy kilku ważnych postulatów.

Ale chciałbym też podziękować za inspirację posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego: za interpelacje, za różne problemy, które były podnoszone, bo z tych refleksji również skorzystaliśmy. Chciałbym również podziękować wszystkim, których nie wymieniłem, za dodatkowe propozycje, za refleksje związane z programem odbudowy i wykorzystaniem środków unijnych.

Szanowni Państwo! To jest chwila, która powinna nas połączyć.

Dzisiaj powinniśmy odłożyć do lamusa wszystkie partykularyzmy partyjne, kalkulacje polityczne niektórych polityków - małostkowe, niepotrzebne. Odłóżmy je na bok. Powinniśmy skupić się na jedności, na zgodzie skierowanej na jak najszybsze wyjście z pandemii, jak najszybszy rozwój Polski, przekazaniu środków dla polskich rodzin, polskich pracowników służby zdrowia, pracowników edukacji, dla Polaków na infrastrukturę w bardzo wielu obszarach. To jest, szanowni państwo, moment arcyważny, moment fundamentalny i w takim fundamentalnym momencie nie ma miejsca na kłótnie, nie ma i nie powinno być miejsca na małostkowe kalkulacje polityczne takie czy inne. Dzisiaj przede wszystkim liczy się Polska. Liczy się interes Polski. To jest przełomowy moment i w takim momencie apeluję do całej Wysokiej Izby o głosowanie za przyjęciem tej ustawy. Ustawy, która tworzy dla nas znakomite, bardzo dobre perspektywy wyjścia z kryzysu. Niech ten przełomowy moment zaowocuje głosowaniem bardzo wielu osób - mam nadzieję, że znacznej większości - za tą ustawą, bo w takim momencie odkładamy na bok kalkulacje, w takim momencie liczy się dobro Rzeczypospolitej, dobro Polaków, liczy się Polska. Dziękuję, panie premierze.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Jak pan premier już powiedział, mamy ważny dzień. W dziejach ojczyzny są chwile niezwykle ważne, gdy dla wspólnego dobra należy odłożyć wewnętrzne spory. Tak było już wielokrotnie - gdy Polska przystępowała do NATO, przystępowała do Unii Europejskiej, być może nieidealnej, na pewno mającej swoje wady, ale jednak będącej projektem bezpiecznej i zasobnej Europy. Możemy być wdzięczni, że w tej Unii jesteśmy. Podobnie też odkładaliśmy takie wewnętrzne spory, kiedy były głosowania zatwierdzające poprzednie perspektywy budżetowe. Były to głosowania niemalże jednogłośne.

Kto wtedy rządził? Też Platforma Obywatelska z PSL-em, Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. Nam nawet do głowy nie przyszło, żeby takim głosowaniem próbować szkodzić Polsce. Byliśmy konstruktywną i odpowiedzialną opozycją. A co mamy dzisiaj? Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki wynegocjował znakomite warunki finansowe nowej perspektywy budżetowej na lata 2021–2027. Fundusz, który ma pomóc gospodarce europejskiej dźwignąć się po dramacie pandemii, ale nie tylko w gospodarce, ma również przygotować służbę zdrowia na ewentualne podobne przypadki.

Tak więc naprawdę jest to znacząca kwota. Są to największe w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej środki dla Polski. W czasie dyskusji było mnóstwo uwag dotyczących samorządów, więc może przeanalizujmy tę kwestię.

Samorządy będą korzystały nie tylko z regionalnych programów operacyjnych, ale jeszcze oczywiście z programów zarządzanych centralnie, bo beneficjentami tych programów centralnych są również samorządy. Dla samorządów są też przewidziane środki z Funduszu Odbudowy - tego specjalnego, na trudny czas w Polsce. Środki z tego funduszu wykorzystywane będą w ramach przygotowanego krajowego programu odbudowy.

A dla przedsiębiorców przewidziano, w formie dotacji, ponad 4 mld euro, czyli blisko 20 mld zł.

Krajowy program odbudowy to jeszcze ochrona środowiska, zmniejszenie energochłonności: ponad 6 mld euro, to transformacja cyfrowa: ponad 3 mld euro, to elektromobilność, energia zielona: ponad 6 mld euro, w tym na sam tabór autobusowy, jak się przyjrzałem, jest ponad 1 mld euro dla samorządów. Kolejna pozycja, czyli ochrona zdrowia: ponad 4 mld euro, w tym dofinansowanie podmiotów leczniczych.

Zapytajmy w powiecie, czy 13 mln to jest dużo czy mało i czy warto z tego skorzystać, czy ważniejsza jest walka polityczna z Prawem i Sprawiedliwością czy jednak możliwość skorzystania z tych środków finansowych.

Właśnie po raz pierwszy jest szansa na uzyskanie średniej europejskiej. Myślę, że nikt się na to nie odważy. Ja tak naprawdę staram się zrozumieć motywy postępowania kierownictwa Platformy Obywatelskiej, jednak przyznaję, że przychodzi mi to z trudem. Słuchałem pana przewodniczącego Borysa Budki, który kilka miesięcy temu wzywał do akceptacji budżetu europejskiego, bez konsultacji, na szybko, ślepo, bez uzgodnień z samorządami, a teraz chce głosować przeciw. Co zatem się zmieniło? Trudno mi jednoznacznie określić, ale pewnie narastająca frustracja z powodu tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości znakomicie sobie radzi w okresie pandemii. Bardzo skuteczna i szybka pomoc przedsiębiorcom w ubiegłym roku spowodowała, że Polska mogła praktycznie, można tak powiedzieć, suchą nogą przejść przez ogromny kryzys. Spadek PKB w 2020 r. był jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej. Bezrobocie praktycznie nie wzrosło, a obecnie jest najniższe w Unii Europejskiej.

Tym, którzy będą głosować przeciw, ludzie nie wybaczą.

Wyczerpał pan czas. Apeluję więc do wszystkich posłów, abyśmy pokazali, że jesteśmy odpowiedzialni za ojczyznę. Jest za co, jest za co. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Borys Budka.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! No cóż, rzeczywiście, przytoczył pan kilka faktów historycznych, kilka dat. Dlaczego tak bardzo atakuje pan ministra sprawiedliwości, koleżanki i kolegów z Solidarnej Polski? Nie potrafił pan przekonać własnego rządu. własnego zaplecza politycznego [[Oklaski]] do decyzji, by poprzeć ratyfikację. Lepiej - kiedy tak naprawdę ważyły się losy Europy, ważyły się losy tego, czy Polska dostanie te fundusze, kiedy w Parlamencie Europejskim zatwierdzano nowe dochody własne, to proszę sobie wyobrazić, co zrobili pana partyjni szefowie: pan Brudziński się wstrzymał, a pani Beata Szydło, pana szefowa, głosowała przeciw. Żaden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w europarlamencie nie poparł decyzji o dochodach własnych. Nikt z was tego nie zrobił. Wówczas szantażowaliście Unię Europejską, szantażowaliście naszych partnerów, atakowaliście wspólne wartości. Dzisiaj zastąpiliście de facto w koalicji rządowej pana Ziobrę, który wyszedł, zwiał, bo chyba nie mógł wytrzymać tych ataków ze strony koalicjantów, nowym koalicjantem - koleżankami i kolegami z Lewicy. To smutne. Bo dzisiaj skończyła się walka o kształt KPO w Sejmie. Ona się nawet nie zaczęła. Ta dezercja i wywieszenie białej flagi spowodowały, że Sejm nie jest miejscem, w którym toczy się merytoryczna debata. Przecież do niedawna cała opozycja mówiła o tym, że Krajowy Plan Odbudowy powinien być dyskutowany tu, w parlamencie. To właśnie w tym miejscu należało upomnieć się o podstawowe zasady, o wartości, które są wspólne dla całej demokratycznej opozycji - uczciwość, sprawiedliwość, jasne, czytelne zasady rozdziału środków europejskich. To właśnie dlatego w 2007 r. i w 2014 r. głosowaliście za tymi dokumentami, o których pan mówił. Bo wówczas gwarantowaliśmy transparentność, uczciwość i przejrzystość tych zasad. Wy zaproponowaliście Polakom, zaproponowaliście polskim samorządom i stronie społecznej całkowitą uznaniowość. Wbrew temu, co mówi wasz nowy koalicjant, w Krajowym Planie Odbudowy nie ma żadnych gwarancji, że samorządy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne będą miały jakikolwiek głos decydujący.

Dzisiaj, wbrew temu, co usiłuje mówić Lewica, w wysłanym do Brukseli Krajowym Planie Odbudowy nie ma żadnej gwarancji, że samorządowcy będą współdecydować o tym, na co zostaną przeznaczone środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma żadnych gwarancji. To jest pierwsze kłamstwo. to nie zaplecze gabinetowe, to nie tajne negocjacje, to nie zakulisowe rozgrywki, to nie pana niemoc we własnym rządzie i próba układania się z częścią opozycji powinny być wyznacznikiem tego, jak działa polski rząd. To właśnie parlament jest miejscem, gdzie trzeba rozmawiać o zasadach, o wartościach, ale przede wszystkim szukać konsensusu. Odrzuciliśmy te wasze zakulisowe gierki, odrzuciliśmy dogadywanie się za plecami innych opozycyjnych partnerów. Krajowy Plan Odbudowy nie mógł podzielić losu funduszu inwestycji lokalnych, ale niestety tak się stało. Stało się tak, dlatego że koledzy, koleżanki z Lewicy uwierzyli panu na słowo. Uwierzyli, że wybudujecie 75 tys. mieszkań, mimo że tego nie ma w KPO. Panie premierze, może pan powie: Gdzie jest te 100 tys. mieszkań? Ile pan wybudował? Wie pan ile? Nawet 2 tys. mieszkań nie potrafił pan przez blisko 6 lat wybudować. Dzisiaj wybuduje pan 75 tys.

O czym od samego początku mówiliśmy? Szanowni państwo, mówiliśmy: tak, te środki Polsce się należą. tylko wam, Polkom i Polakom, którzy tak ciężko znieśliście kryzys gospodarczy. Należą się wam, którzy dzielnie walczycie, wbrew temu nieudolnemu rządowi, z pandemią. Proponowaliśmy wielki plan zdrowia dla Polaków. Proponowaliśmy konkretne rozwiązania. A co zamiast tego mamy? Zamiast tego jest tajny plan, którego nawet nie widziała komisja trójstronna. Tajny plan, którego nie zaakceptowała strona samorządowa. Dzisiaj, kiedy słyszę z ust koleżanek i kolegów z Lewicy, że mówią w imieniu samorządów, to ja chcę zerknąć np. na waszą przedstawicielkę w komisji wspólnej, w Związku Miast Polskich. Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która w sojuszu Lewicy jest od 2014 r., mówi wyraźnie: nawet z nią nie konsultowaliście waszych propozycji. A dlaczego? Dzisiaj w Senacie odbyliśmy szybkie wysłuchanie publiczne z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządu. Prosili o czas. Prosili o to, żeby mieli możliwość wynegocjowania dobrych warunków z rządem. Tymczasem do czego wy doprowadziliście? Zmusiliście rząd, żeby wysłał nikomu nieznany dokument przed zakończeniem negocjacji z samorządowcami. Na Boga, koleżanki i koledzy, tak się nie robi. Dzisiaj zostawiliście nie tylko opozycję - bo to rozumiem, możemy się różnić - ale zostawiliście organizacje pozarządowe, zostawiliście samorządowców. Zostawiliście ich na spalonych. Ja słyszę: dlaczego. Naprawdę, koleżanki i koledzy, wy dzisiaj myślicie o tym, żeby się ścigać w opozycji? O jakichś liderach opozycji? To ja wam przypomnę, że już jeden lider opozycji siedział na waszych miejscach. Jak skończył w tym wyścigu, to wszyscy wiemy. Dzisiaj jest wielkie wyzwanie dla całej opozycji. Dzisiaj jest czas na to, by współdziałać, a nie dzielić. Dzisiaj jest czas na to, by pokazać, że rząd nie ma większości, by zmusić do tego, by Krajowy Plan Odbudowy był rzetelnym dokumentem, który uzyska konsensus społeczny. Była szansa na to, by zmusić rząd do rozmów w parlamencie. Niestety wy jej nie wykorzystaliście. Dlatego chcę raz jeszcze podkreślić: od samego początku byliśmy za tym, żeby do Polski trafiły te pieniądze. Wszyscy eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, zarówno nasi przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i z Platformy Obywatelskiej, głosowali za tymi pieniędzmi dla Polski. Jednocześnie żądaliśmy transparentności, uczciwości, ale przede wszystkim tego, by 40% środków, tak jak do tej pory, było rozdzielane przez samorządy. Dzisiaj zgłosiliśmy szereg poprawek. Nawet tych poprawek nasi przyjaciele z opozycji nie byli w stanie poprzeć, nawet gwarancji 40% środków właśnie dla samorządów. Mówię o tej stronie opozycji. Ale jest jeszcze czas na to, by to poprzeć w Senacie. Dzisiaj to nie jest miejsce do tego, by rozgrywać jakieś partyjne interesy. Dzisiaj parlament powinien być miejscem, gdzie w konsensusie zatwierdzimy dobre decyzje dla Polaków. Wybraliście inną drogę.

Dlaczego? Bo nie upomnieliście się o wartości. Zostawiliście Polki, które na ulicach obrywały pałami od tego rządu. Woleliście zakulisowe rozgrywki. Wróćcie na dobrą stronę opozycyjną. Jest jeszcze czas. Zgłaszamy (Dzwonek), panie marszałku, szereg poprawek w drugim czytaniu. Jednocześnie deklaruję, że nie będziemy popierać tego rządu. Wstrzymamy się, jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte. Ale jest szansa, by dzięki tym poprawkom zagwarantować uczciwy plan odbudowy, zagwarantować fundusze dla samorządów, komitet monitorujący, ale przede wszystkim zagwarantować transparentność i sprawiedliwość tych środków. Nie mogą podzielić środków, które zostały wyrzucone w błoto, na wasze inwestycje w Ostrołęce, na Centralny Port Komunikacyjny, na propagandę w państwowej telewizji, na zakup prywatnych mediów dla celów propagandowych. Te propozycje gwarantują, że będziemy wam patrzeć na ręce.

Panie pośle, różne dziwne rzeczy pan tu opowiadał, ale jedno muszę sprostować w imieniu naszych nieobecnych kolegów. Nasi parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim głosowali za tym projektem, a w drugim głosowaniu, dotyczącym długu, cztery osoby głosowały przeciw, natomiast miażdżąca większość, 23 osoby, głosowała za. Bardzo proszę, teraz w imieniu Lewicy pan poseł Adrian Zandberg.

Wysoka Izbo! Mój poprzednik przez 10 minut zamiast o Funduszu Odbudowy opowiadał o tym, jak bardzo nie podoba mu się Lewica. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy skupili się na rzeczach ważnych. To był zły rok dla Europy. Epidemia zabiła setki tysięcy z nas i zrujnowała życie milionom. Od Warszawy po Madryt, od Kopenhagi po Ateny - wszędzie czekamy na powrót do normalności. Ci, którzy nieśli pomoc, i ci, którzy tej pomocy potrzebowali. Ci, którzy potracili bliskich, i ci, którym udało się uchronić przed wirusem. Ten zły rok wstrząsnął Europą. Wierzę głęboko, że możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi. Po to jest ten wielki plan, żeby postawić Europę na nogi po epidemii, żeby ruszyć do przodu, żeby wybrać przyszłość. I o tym dzisiaj warto rozmawiać, bo już za chwilę w tym głosowaniu będziemy decydować w imieniu Rzeczypospolitej o pogłębieniu integracji europejskiej. Jeżeli powstanie Europejski Fundusz Odbudowy, to zapewnimy miliardy euro dla Polski i uczynimy Unię silniejszą i bardziej zjednoczoną. Jeżeli jednak fundusz upadnie, to będzie zwycięstwo wrogów Europy, obecnych niestety także tutaj, na tej sali, bo ci, którzy chcą zniszczyć Unię, marzą o tym, żeby fundusz upadł, bo wiedzą, że w ślad za tym rozpadnie się nadzieja na silną Europę. I to jest prawdziwa stawka tego głosowania. Kto zagłosuje dzisiaj za ratyfikacją, głosuje za silną Europą, a ten, kto nie umie podnieść ręki za ratyfikacją, głosuje za Europą słabą, za Europą bezsilną, za Europą bezbronną. Dzisiaj bloki gospodarcze na całym świecie uruchamiają inwestycje. Stany Zjednoczone prezydenta Bidena ruszyły do przodu. Tak samo robią Chiny. Europa nie może zostać w blokach startowych. Europejski Fundusz Odbudowy to są wielkie publiczne inwestycje, to są pieniądze na ratowanie miejsc pracy, to są pieniądze na kolejne oczyszczalnie ścieków, na panele fotowoltaiczne i na farmy wiatrowe, na mieszkania dla młodych, na finansowanie badań naukowych, na kształcenie lekarzy, na robotyzację przemysłu, na sieć piątej generacji, na technologie wodorowe, na magazyny energii, na nowoczesną gospodarkę. To jest szansa na skok cywilizacyjny.

Ale nie jest niestety powiedziane, że w tym wielkim projekcie wezmą udział wszyscy. Już raz Polska nie wzięła udziału w planie Marshalla. Do dziś płacimy za to cenę. Jeśli Polska nowy plan Marshalla odrzuci, mniejsza o to, z jakich przyczyn, to Zachód po raz kolejny nam ucieknie. Tym razem na szczęście nikt nie decyduje za nas. Wszystko jest tu, w tej sali, w naszych polskich rękach. I przypominam to wszystkim, którzy będą głosować na tej sali, bo nie wolno raz jeszcze popełnić tego samego błędu. Mówiłem o pandemii, ale pandemia to nie jest jedyne wyzwanie przed Europą. Musimy zatrzymać zmiany klimatu. Są oczywiście na tej sali politycy nieodpowiedzialni, tacy, którzy udają, że kryzysu klimatycznego nie ma. Ale każdy rok bezczynności spycha naszą planetę na krawędź dramatycznego kryzysu, na krawędź katastrofy. Musimy podnieść efektywność energetyczną. To oznacza, że musimy odejść od paliw kopalnych. Europejski Fundusz Odbudowy to są środki na zieloną transformację. Potrzebujemy tych pieniędzy. Europejskie gospodarki, w tym gospodarka polska, muszą stać się neutralne klimatycznie, bo jeżeli nie zrobimy tego na czas, to świat, w którym będą żyły nasze dzieci, po prostu stanie w płomieniach. Wysadzenie w powietrze Europejskiego Funduszu Odbudowy to jest wysadzenie w powietrze przyszłości naszych dzieci i wnuków, to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Słyszę, że pan minister Ziobro mówił dzisiaj w Sejmie, że będzie głosować przeciwko, bo ten fundusz to jest federalizacja Europy, to jest krok w stronę europejskiego superpaństwa. Odpowiadam panu ministrowi Ziobro. Nie myli się pan, panie ministrze. I bardzo dobrze, że tak jest, bo nowe wspólne inwestycje publiczne zwiążą nas silniej z Europą. a europejski mechanizm praworządności utrudni panu, panie ministrze, bezkarne niszczenie polskich sądów. Przyznaję, panie ministrze Ziobro, że panu ta ratyfikacja musi być wyjątkowo nie w smak. Europa, szanowni państwo, to jest polska racja stanu. Europa to jest najlepsza gwarancja demokracji i praworządności. Chciałbym, żeby ci, którym chodzi dziś po głowie rozwalanie funduszu w imię partyjniackich gierek, byli świadomi konsekwencji, bo europejski pociąg może odjechać bez nas. W Berlinie, Paryżu, Amsterdamie są politycy, którzy myślą, że może łatwiej byłoby bez Polski. Po jednej stronie jednocząca się Europa, po drugiej stronie agresywna Rosja, a w środku my, pozbawieni europejskich funduszy i odcięci od Zachodu. To jest najgroźniejszy scenariusz dla Polski. To jest scenariusz, do którego nie wolno dopuścić. My, Lewica, chcemy Europy silnej, ale wiemy, że sama siła nie wystarczy, bo każdy łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego Europa musi być solidarna. Nie zostawiamy w potrzebie tych, którym wiedzie się gorzej. Wspólne europejskie zadłużenie to jest solidarność w działaniu. I ta europejska solidarność nie może kończyć się na poziomie państw. Musimy zadbać o ludzi. Pieniądze są po to, żeby rozwiązywać ich problemy, żeby pomóc tym, którzy są w potrzebie. I o to walczyła Lewica w trakcie negocjacji, o zdrowie, o mieszkania dla młodych, o ratowanie miejsc pracy. Mam nadzieję, że po roku pandemii już wszyscy na tej sali, także w tej części sali, zrozumieli, że potrzebujemy silnej publicznej ochrony zdrowia, bo w Polsce umarło 100 tys. ludzi na darmo, ludzi, którzy mogli żyć.

Szpitale muszą być lepiej dofinansowane i muszą one być lepiej dofinansowane wszędzie.

I zapewniliśmy środki dla szpitali powiatowych. Musimy wreszcie zadbać o młodych. To jest problem numer jeden tego pokolenia - mieszkania. Było wiele hucznych zapowiedzi w Polsce, na tej sali, ale nigdy nie poszły za tym konkretne pieniądze. Teraz jest szansa, żeby to zmienić. Dlatego wymogliśmy wpisanie mieszkań do Krajowego Planu Odbudowy. Niektórzy powiedzą, że te dziesiątki tysięcy mieszkań to jest kropla w morzu potrzeb. I ja się zgadzam, macie rację, bo prawdziwą zmianę oczywiście przyniesie dopiero lewicowy rząd, ale każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku i to jest właśnie ten pierwszy krok.

Przy centralnych ulicach dużych polskich miast i małych miasteczek straszą poopuszczane lokale, puste knajpy. Te miejsca trzeba ożywić. Trzeba odtworzyć te miejsca pracy. Trzeba pomóc im stanąć na nogi. Lewica walczyła o pomoc dla tych ludzi i ta pomoc będzie, europejskie środki na to będą z Europejskiego Funduszu Odbudowy. My w Lewicy tak właśnie rozumiemy politykę. Jesteśmy w parlamencie po to, żeby walczyć o sprawy zwykłych ludzi. Innym zostawiamy rojenia o księżycowych koalicjach z panem Braunem i z panem Bosakiem. Te miliardy euro będą dla Polski pomocą i zastrzykiem energii, bez którego polska gospodarka może sobie nie poradzić. Obowiązkiem odpowiedzialnych polityków jest te pieniądze Polsce zapewnić. Wysoka Izbo! Rządy przychodzą i odchodzą, także te złe rządy, takie jak ten, który rządzi dziś Polską, ale zostaje Polska. I dziś decydujemy o przyszłości naszego kraju i o przyszłości Europy. Konsekwencje tych głosowań zostaną z nami na lata. Będzie się z nimi mierzyć nie tylko ten rząd, ale wszystkie kolejne rządy. Warto być świadomym wagi tych rozstrzygnięć. Europa to jest polska racja stanu. Lewica zagłosuje za Europą, Lewica zagłosuje za polską racją stanu. Zapraszam do zabrania głosu pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza, Koalicja Polska. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Zrzuciłem garnitur, założyłem fartuch i ostatnie tygodnie spędziłem w izbie przyjęć krakowskiego szpitala na pierwszej linii frontu walki z COVID-em.

Ale są one potrzebne rzetelnie i transparentnie podzielone. Dla wszystkich, nie dla wybranych, nie dla samych swoich, tak jak Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dlatego od początku dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy i Funduszu Odbudowy stawialiśmy warunki - jako pierwsze ugrupowanie, później dołączyły kolejne, za co bardzo dziękuję. Stawialiśmy warunki dotyczące udziału samorządu, udziału przedsiębiorców prywatnych, żeby nie była to jakaś gigantomania ani megalomania na wzór Gierka, którego długi spłacaliśmy przez kolejne dziesięciolecia. Chodzi o to, żeby te pieniądze trafiły do wszystkich wspólnot lokalnych, do wszystkich samorządów, niezależnie od koloru legitymacji partyjnych włodarzy gmin, powiatów i województw.

Historycznie Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój wielki udział w przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pan premier mówił o tej historii, ale o tym nie wspomniał, więc ja naprostuję i rozjaśnię. To Jarosław Kalinowski heroicznie negocjował najlepsze możliwe warunki dla polskiego rolnictwa, a później razem z Platformą negocjowaliśmy najwyższy historyczny budżet z Unii Europejskiej. I to są rzeczy, które dają nam świadectwo bycia zawsze za Europą, za silną Polską w Europie, za pogłębioną integracją. Pan premier szukał przed chwilą przeciwników Funduszu Odbudowy w Europie. Panie Premierze! Najpierw trzeba w swojej zagrodzie przekonać trzódkę Solidarnej Polski. Bliżej trzeba spojrzeć, gdzie są ci przeciwnicy. Oni siedzą razem z panem w ławach rządowych. Oni od początku panu mówią, że jest pan zdrajcą, że to jest utrata suwerenności. To jest poważna sprawa. A pan mówi dzisiaj: to jest miara naszego patriotyzmu - bycie w Unii i skorzystanie z tych pieniędzy. Chce pan przekonać opozycję i słusznie, bo to jest pana obowiązek budować większość w odniesieniu do swoich projektów, ale zawsze trzeba zacząć od tych, którzy z panem od 5 lat współrządzą. To się nie udało i to jest gigantyczna porażka. Teraz o polityce, o której było dużo w wymianie zdań miedzy Lewicą i Platformą. Niedobrze, że do tego doszło. W pewnym momencie mieliśmy solidarność, razem organizowaliśmy wysłuchanie publiczne, mieliśmy wspólne postulaty, dla nas bardzo ważne, dotyczące rolnictwa, dotyczące polskiej wsi, rzemiosła, przedsiębiorców, dla Lewicy np. dotyczące spółdzielców, w przypadku Platformy - wspólnot lokalnych, również samorządowców. Dla nas wszystkich to były ważne tematy i gdybyśmy tę jedność utrzymali do końca, wynegocjowalibyśmy dużo więcej. Moglibyśmy pomóc naprawdę na transparentnych, jasnych zasadach wszystkim, a nie tylko małej grupie. Szkoda, że tę solidarność w opozycji utraciliśmy. I wiecie, kto się z tego najbardziej cieszy? Prezes Jarosław Kaczyński i prezes Zbigniew Ziobro.

Niestety, bo moglibyśmy przedstawiać dzisiaj Krajowy Plan Odbudowy na zasadach wspólnot lokalnych, samorządowców, NGO i przedsiębiorców. Trochę rzeczy się udało i też chcę oddać prawdę. Początek był fatalny, panie premierze. Zaczęliście od Krajowego Planu Odbudowy, w którym było 250 stron, ale tak naprawdę nic z niego nie wynikało. Nie było tam strategii, myśli.

Powołanie komitetu monitorującego samorządowców, złożonego z samorządowców i organizacji pozarządowych i 1 mld zł na inwestycje w zeroemisyjny transport szynowy. To np. dla Warszawy, dla mojego rodzinnego Krakowa jest bardzo ważne. Wiem, że też pan prof. Majchrowski składał takie postulaty. Nie udało się też zmienić wymiaru sprawiedliwości, bo przecież w krajowym planie są też intencje zmian systemowych. Gdybyśmy do końca negocjowali wspólnie, do ostatniego dnia, dopóki jest to możliwe i nie pokazali wszystkich kart, jak chcemy zagłosować, transparentność i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jego niezawisłość i niezależność byłyby większe. Niewystarczająco został wzmocniony też fundusz spółdzielczy. To, co się udało osiągnąć, również naszemu klubowi, Koalicji Polskiej - PSL, zawdzięczamy tym, którzy brali udział w konsultacjach - samorządowcom wszystkich szczebli, wszystkim organizacjom pozarządowym. Szczególnie dziękuję Kubie Wygnańskiemu za zorganizowanie prawdziwej debaty, burzy mózgów nad tym wszystkim, co się dzieje z krajowym planem, z Funduszem Odbudowy. Nie jakakolwiek partia polityczna, nie ta po lewej czy ta po prawej, czy nawet ta pośrodku. Prawdziwym zwycięzcą tego wszystkiego muszą być kolejne pokolenia. Musimy się podnieść nie tylko w momencie zapaści epidemiologicznej, ale musimy się podnieść z zapaści. w którą czasem sami się wprowadzamy przez przeregulowanie gospodarki, tysiące stron ustaw, które są produkowane, biurokratyzację, która zaczyna nas zżerać, co też dobrze widać w szpitalach. Dzisiaj będziemy podejmować decyzje - i od naszego głosu, naszego klubu bardzo dużo zależy - jak zagłosujemy, jak to będzie wyglądać. Chcemy mieć też gwarancję, dlatego zgłaszamy poprawki, żeby ten fundusz był dobrze wydatkowany. W 18. roku naszej obecności w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy spowodowany pandemią. Rzeczpospolita Polska, ratyfikując Fundusz Odbudowy, potwierdza, że jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest solidarność europejska. Władze Rzeczypospolitej zobowiązują się, że środki będą wydatkowane na zasadach sprawiedliwych, transparentnych, opartych na wartościach demokratycznego państwa prawa. rolników, organizacji pozarządowych, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Środki z Funduszu Odbudowy mają służyć modernizacji państwa, rozwojowi innowacyjności, gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Kto za tym nie zagłosuje, ten będzie chciał coś chachmęcić, ten będzie chciał rozdawać te środki w nieprawidłowy sposób. To jest poprawka dotycząca zasad praworządności, zasad zgodności z konstytucją, z prawem europejskim.

To są gwarancje rzetelności wydatkowania tych środków i one powinny być zapisane w ustawie, nie tylko pozostać jako deklaracje słowne. Dzisiaj nie zagłosujemy razem z kimś. Dzisiaj nie zagłosujemy za rządem.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Bosak, proszę.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka, ale coraz niższa Izbo! Dzisiejsze posiedzenie to jest Sejm rozbiorowy. Dzisiaj zdecydujemy o tym, czy Polska odda się w jeszcze głębszą niewolę Brukseli, czy za paciorki sprzeda kolejny kawałek swojej suwerenności. Posłowie z prawej strony, którzy macie zamiar podnieść za tym rękę, mam prośbę: odwróćcie te swoje przypinki w klapach do góry nogami. Nie szargajcie symboli, które zaraz będziecie zdradzać. Może jesteście patriotami z Indonezji, ale na pewno nie z Polski, tak że bardzo bym o to prosił. Jesteście tak naprawdę tylko kacykami uganiającymi się za doraźnymi korzyściami, za doraźnymi pieniędzmi na przekupywanie wyborców, byle jakoś dojechać do kolejnych wyborów. I tak jak plemienni kacykowie sprzedawali swoich ludzi w niewolę za paciorki, żeby chwilowo skorzystać z doraźnych korzyści, jakie te paciorki im na miejscu dawały, tak wy nas sprzedajecie za 600 euro od głowy pod dyktat obłąkanego imperium brukselsko-berlińskiego pod tęczową flagą. Zostaliście wybrani po to, żeby strzec suwerenności, a rozmieniacie ją na drobne. Robicie dokładnie to, co zrobiłaby na waszym miejscu Platforma, więc co za różnica. Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników, różnica jest taka, że wy weźmiecie więcej. Ale mam nadzieję, że tak samo udławicie tymi pieniędzmi. Naprawdę trudno mi uwierzyć, że nie widzicie konsekwencji, że na tej politycznej planszy nie potraficie przewidzieć dwóch ruchów do przodu. Pozwalacie obcej organizacji ściągać trybut z terytorium Rzeczypospolitej, taki jaki ona uzna za stosowny. To ja się pytam, jaką my wojnę przegraliśmy, że się na coś takiego musimy zgadzać. Może gdybyście przez poprzedni rok nie bombardowali własnego terytorium, swoimi durnymi ustawami nie zadławili gospodarki, to teraz nie musielibyście sprzedawać nerki, żeby się ratować. Pan premier nawiązał tutaj do planu Marshalla.

Bo Niemcy postawili na niskie podatki i wolny rynek, a nie na rozdawnictwo pożyczonych pieniędzy. To są pieniądze, które zostaną wydarte obywatelom, żeby napchać kieszenie banksterów. I tutaj kłaniam się w lewą stronę. Bierzecie po raz kolejny państwo udział w transferze pieniędzy od biednych do bogatych. To klasa robotnicza będzie wydawała te pieniądze rękami swoich najznakomitszych przedstawicieli w Warszawie, a banksterzy już zacierają ręce, nie mogą się doczekać odsetek, które przez pokolenia będą spłacane, bo państwa nie spłacają długów, tylko je rolują w nieskończoność. Zastanówcie się, co robicie.

Proszę bardzo, dokończy pan poseł Krzysztof Bosak. Szanowni Państwo! Być może ktoś, słuchając tej debaty, zastanawia się, dlaczego premier Morawiecki mówił tak bardzo bez przekonania, dlaczego minister Kowalczyk mówił tak bardzo bezbarwnie i dlaczego Adrian Zandberg tak świetnie dziś czuł się na mównicy, mówił z takim przekonaniem. Z bardzo prostego powodu: dziś Lewica realizuje swój program i może być z tego dumna. Mówi o tym otwarcie, nie wprowadza opinii w błąd. Mówi: wzmacniamy Unię Europejską, posuwamy integrację unijną do przodu. Zaś to, co robi PiS, to próba ukrycia przed opinią publiczną tego, co rzeczywiście robicie. Pan premier Mateusz Morawiecki, były doradca premiera Donalda Tuska, wie najlepiej, co robi. Lewica realizuje swój program. Z prostego powodu. Dziś głosujemy dlatego, że przesuwamy nowe kompetencje do Brukseli. Teraz przejdzie. Bruksela będzie wyliczać, na co da temu i przyszłym rządom pieniądze.

Wejdą nowe podatki unijne, o których nikt nie wspomniał: od plastiku, od śladu węglowego, cyfrowy, od transakcji finansowych. PiS zdradził polskich patriotów, umacnia Unię Europejską, a nie Polskę.

Wysoka Izbo!

Jaki świat im zostawimy? Czy będą mogli w nim spełniać swoje marzenia? To, jaką Polskę i Europę przekażemy naszym dzieciom, decyduje się dzisiaj, tu i teraz. Dlatego Polska 2050 jako jedyna niezmiennie i konsekwentnie opowiada się za jego przyjęciem. Do egzaminów dojrzałości przystępujemy dzisiaj jako cała klasa polityczna. Niektórzy z nas siedzą tu z dzienniczkiem pełnym uwag i trudno mieć do nich zaufanie. Niektórzy nadal wahają się, czy nie postawić rządowi jedynki. Ale nadal wszyscy mamy szansę dzisiaj zdać ten test. Nie dla rządu, a pomimo niego.

Proszę. Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Fundusz Odbudowy to sprawa zbyt poważna, by nadal mogła być pretekstem do wymiany wzajemnych złośliwości i popisywania się przez polityków arogancją. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni takim stylem uprawiania polityki, a Polacy od wielu tygodni nie rozumieją tego, co do nich mówicie. Obywatele oczekują od nas przede wszystkim dojrzałości, zwłaszcza gdy mówimy o pieniądzach, które powinny stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki na kolejną dekadę. Ubiegły rok zamknęliśmy deficytem na poziomie 161 mld zł. Każdego dnia ludzie tracą swoich bliskich. Pieniędzy, których żaden europejski rząd nie ma prawa upolityczniać, również wy, panie premierze. To nie są pieniądze partyjne, premierze Morawiecki. To nigdy nie były i nigdy nie będą wasze pieniądze. To są pieniądze obywateli Europy. I na tych pięknych lawetach dobrze by było wyraźnie pokazać flagę Unii Europejskiej, panie premierze. Fakt, że nie zorganizowaliście w Sejmie debaty nad ostatecznym kształtem Krajowego Planu Odbudowy przed jego wysłaniem do Brukseli, jest dowodem na małość i partyjniactwo, które uprawiacie. Miejsce debaty nad Krajowym Planem Odbudowy jest tutaj, w Sejmie, na sali plenarnej, a nie w gabinetach klubowych czy ministerialnych. Nasze stanowisko jest niezbędne. Część z nich podzieliła Komisja Europejska, choć panu premierowi Morawieckiemu do dziś słowo Polska 2050 nie przechodzi przez gardło. Tak, złożyliśmy je, panie premierze, 17 marca. Oczywiście jest wiele do dopracowania, m.in. mechanizm kontroli. Unia musi dowieźć ten plan. Unia musi być silna i solidarna, zjednoczona, musi pogłębiać współpracę o kolejne obszary, zwłaszcza w dobie nasilających się kryzysów na Wschodzie. Słaba Unia to większa przestrzeń dla takich ludzi jak Zbigniew Ziobro, przestrzeń do niszczenia niezależnych instytucji demokratycznego państwa prawa. Nie przyłożymy do tego ręki. Nie będziemy mówić głosem Zbigniewa Ziobry czy konfederatów. Czy mamy obawy, że PiS będzie chciał upolityczniać te pieniądze i dawać je swoim? Oczywiście, że mamy, ale widzimy, że Komisja Europejska wyciąga wnioski z ostatnich lat i wie, że musi zadbać o rzetelne i transparentne wydatkowanie pieniędzy. Krajowy Plan Odbudowy to nie jest zwykła formalność, którą klepniecie sobie na Nowogrodzkiej. Ma być twardą podstawą do oceny, czy rząd będzie wydawać te pieniądze zgodnie z unijnymi celami. Premierze Morawiecki, do przegranych wyborów zostało panu 2 lata. Przez ten czas będziemy patrzeć wam na ręce.

Wysoka Izbo! W imieniu koła Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące druku nr 1123 o ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Na wstępie pragnę zauważyć, iż gospodarki wielu państw ucierpiały wskutek licznych lockdownów stosowanych w ostatnim roku, jak również wskutek zerwania łańcuchów dostaw i powstałej w wyniku tego paniki. Fundusz Odbudowy i związany z nim Krajowy Plan Odbudowy nie powinny być elementem bieżącej gry politycznej, ale głębokiej refleksji zgodnej z polską racją stanu. Wielu Polaków liczy na te pieniądze, bo chcą wyrwać się z wieloletniej biedy i przepaści między Polską a starymi krajami Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, iż są to duże pieniądze, które mogą znacząco wpłynąć na stan naszej gospodarki i dobrobyt Polaków pod warunkiem, iż będą wydane na inwestycje, a nie na bieżące łatanie dziur budżetowych, jak to już wielokrotnie miało miejsce od 2004 r. Z drugiej strony wiemy, iż nie ma darmowych obiadów, za wszystko trzeba płacić. Dlatego tak ważne są szczegóły tego unijnego porozumienia, a dokładnie sposób jego spłaty. Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź na moją interpelację nr 21581, za którą ministrowi Waldemarowi Budzie dziękuję. Pragnę zwrócić uwagę na bardzo niepokojące informacje przekazane przez pana ministra. Problem, który zauważam, a którym nie interesuje się żadne inne ugrupowanie, to sposób spłaty otrzymanych pieniędzy, bo obecnie pieniądze, które mają być pozyskane w ramach Funduszu Odbudowy, wyglądają jak chwilówka, nie znamy szczegółów spłaty. To jakby rodzina robiła gigantyczne zakupy na kredyt, nie zastanawiając się nad tym, jak w przyszłości te pieniądze spłaci. Obawiam się, czy nie będzie tak, jak z pseudokredytami frankowymi, przez które wiele polskich rodzin popadło w niespłacalne długi. Na podstawie odpowiedzi pana ministra obecnie nie wiemy, jaki będzie koszt pozyskania pieniędzy przez Komisję Europejską, nie wiemy, jak będą wyglądały podatki, z których będą następnie spłacane pozyskane środki, i czy rząd obniży podatki krajowe w związku z nowymi podatkami unijnymi, aby nie dokładać dodatkowych obciążeń Polakom, czyli nie znamy najważniejszej kwestii przy zaciąganiu długu. Ile to będzie nas kosztowało? Idąc do banku, pytamy o RSO, czyli całkowity koszt pożyczki. Tutaj, zgodnie z odpowiedzią pana ministra, jest on nieznany. Są to obecnie kluczowe kwestie, gdyż politycy powinni patrzeć dalej niż do najbliższego sondażu czy najbliższych wyborów. Zadłużamy nasze dzieci i wnuki, dlatego powinniśmy wiedzieć, ile pieniędzy będą nasi potomkowie spłacali. Nie mogę odnieść się do peanów wznoszonych przez posłów Lewicy na cześć głębszej integracji europejskiej. Jeżeli wynegocjowane porozumienie rzeczywiście oznacza pogłębioną integrację, nakładanie nowych podatków, groźbę spłacania długów innych państw oraz federalizację Unii Europejskiej, to w tej sprawie powinno odbyć się referendum ogólnokrajowe, bo wszyscy Polacy powinni decydować o tym, jak daleko chcą być zintegrowani w ramach Unii Europejskiej oraz ile suwerenności chcą oddać urzędnikom brukselskim. Dlatego ponownie zapytam pana ministra, pana premiera: Czy to porozumienie oznacza głębszą integrację europejską wraz z wymienionymi konsekwencjami? Kolejna kwestia, którą chcę poruszyć, to aspekt wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi właściwie o tę część skierowaną na wieś i obszary wiejskie. Na obszarach wiejskich mieszka 40% Polaków. To również ponad 90% obszaru Polski. Obszary te od lat były zapomniane i zaniedbane. Mieliśmy zamykane ośrodki zdrowia, komisariaty, poczty. Na obszarach wiejskich jest bardzo dużo miejsc bez Internetu, dostępu do gazu, kanalizacji czy komunikacji masowej. Spłacać Fundusz Odbudowy będzie całe polskie społeczeństwo. Stąd moje kolejne pytanie, na które nie uzyskałem dotychczas odpowiedzi: Jaki całościowy procent środków z Funduszu Odbudowy będzie skierowany na obszary wiejskie według szacunków rządu? Gdyż w mojej ocenie tereny wiejskie zasługują na środki odpowiadające procentowi społeczeństwa zamieszkującego te obszary. Uprzejmie proszę pana premiera o merytoryczne odpowiedzi i przekonanie posłów Kukiz’15, iż te środki będą służyły Polakom (Dzwonek), a nie staną się funduszem wyborczym. Wysoki Sejmie!

Dziękuję, panie pośle. Zapraszam do zabrania głosu panią poseł Agnieszkę Ścigaj, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Proszę. Wysoka Izbo! Po pierwsze, jeśli chodzi o warunki finansowe krajowego programu odbudowy, czyli te związane ze wspólnym kredytem, wspólnymi zobowiązaniami, wspólnymi podatkami, one tak naprawdę zostały już ustalone w grudniu.

Takie są fakty. Możemy mieć uwagi co do sposobu wydawania tych środków, o tym za chwilę, natomiast ważny jest też sposób procedowania, o którym chcę wspomnieć i na który chcę zwrócić uwagę. Organizacje pozarządowe wykonały gigantyczną pracę, przeprowadzając konsultacje społeczne, przeprowadzając tak naprawdę wysłuchanie publiczne, które powinien zrobić rząd. Teraz proszą o to, aby dać im jeszcze tydzień albo dwa, żeby zorganizować odwrócone wysłuchanie, żeby rząd odpowiedział na pytania. Rząd nie szanuje posłów, parlamentarzystów, dlatego że ta dzisiejsza debata trochę mija się z celem, skoro program został wysłany, ale warto wykazać się szacunkiem dla organizacji pozarządowych, dla partnerów, których zaprosiliście do współpracy w komisji trójstronnej. Powołaliście zespół. Zespół pracuje, ma pracować nad ustawą wdrożeniową, bo ona jest kluczowa. Warto znać założenia tej ustawy, panie premierze, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy będzie przejrzystość, jak te środki będą dysponowane, czy w komitecie monitorującym znajdzie się miejsce dla organizacji pozarządowych. Dlatego ze względu na nich, na tych partnerów, trzeba odłożyć to głosowanie o tydzień. Mamy odbudować polską gospodarkę. Przedsiębiorcy. Prawie 2 mln ma problemy, a 500 tys. już zamknęło swoją działalność.

To one się wzmacniały. Ubezpieczenia dla polskich firm, kredyty, gwarancje, zwolnienia podatkowe, zamówienia publiczne, które pozwolą, jak w innych krajach, mieć pierwszeństwo polskim firmom. Czy znowu będziemy tylko takim transferem tych środków unijnych? Druga sprawa.

W tej chwili mamy 500 tys., również za sprawą dystrybucji środków unijnych. Przecież naprawdę mamy dużo urzędów i instytucji. Czy nie lepiej je zaangażować, a nie tylko powoływać ciągle nowe? Mamy jakieś branżowe centra kompetencji, mamy Agencję Rozwoju Szpitali, centra doradztwa i poradnictwa, centra technologii wodorowych. Tego tutaj nie wymienię, ale naprawdę jest dużo, dużo instytucji. Polskie Sprawy pytają w imieniu przedsiębiorców: Czy skoro tak mało środków do nich trafi, a to oni będą musieli wyciągać gospodarkę z kryzysu, rząd planuje rzeczywiście pomóc im w tym, aby te pieniądze również pośrednio u nich zostały? Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Stajemy dzisiaj rzeczywiście przed bardzo trudną, szekspirowską sytuacją. Z jednej strony oczywiste jest, że pieniądze dla ochrony zdrowia są potrzebne i ten resort ciągle wymaga zasilenia. Ale z drugiej strony problem jest też w tym, czy sensownie i dobrze te pieniądze wydamy. Bo wydajemy zwiększone środki już od wielu lat i z tego nic dla pacjentów tak naprawdę nie wynika. Czy państwo słyszeliście, żeby w czasie COVID-u, ale i wcześniej głównym problemem ochrony zdrowia były problemy strukturalne? Nie.

Niestety plan odbudowy przewiduje przede wszystkim wydanie pieniędzy na strukturę, na kolejne inwestycje.

Funkcjonuje lepiej? Testy. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Bardzo ucieszyła mnie decyzja rządu o odmrożeniu kultury, bo chciałem wybrać się

Gospodarka płonie.

A wy tak się zapędziliście w tej plemiennej wojnie, w tym podziale Polaków na Hutu i Tutsi, że zaślepieni nienawiścią do Jarosława Kaczyńskiego chcecie dokonać rytualnego mordu na polskich przedsiębiorcach. Panie Budka, pan został już grabarzem Platformy, a teraz chce pan zostać chyba grabarzem Polski.

I teraz, kiedy Lewica podjęła tę propolską, dobrą i odpowiedzialną decyzję, pan się tak zakiwał i próbuje zakiwać całą opinię publiczną, że wyleciał pan poza boisko wytyczone przez linię logiki, zdrowego rozsądku i polskiej racji stanu. Skala absurdu jest tak duża przy całej dyskusji nad KPO, że gdyby przy jednym stole posadzić Hitchcocka, Mrożka i Bareję, postawić na tym stole 3 l dobrego polskiego rasowego alkoholu, to myślę, że egzotyka intelektualna nie byłaby tak duża jak przy tej dyskusji.

Ale nie można śmiać się z pomylenia interesu Polski z interesem Platformy i chęci ugrania kilku punktów politycznych tylko na tym, żeby zrobić na złość PiS-owi. Tylko że wy nie robicie na złość PiS-owi.

Ta walka plemienna zaszła tak daleko, że mam wrażenie, że jak PiS złoży ustawę o tym, że Ziemia jest okrągła, to pan zagłosuje przeciw tylko po to, żeby zrobić na złość.

Ale to zwykłe wkładanie kija w szprychy sprawia, że właśnie dzięki takim działaniom największy opozycyjny okręt na polskiej scenie politycznej spod bandery Platformy został zredukowany do pozycji wraka. Okej. Panie premierze, ja też nie kupuję działań rządu w całości, sorry.

Zero. Bo, panie przewodniczący, troska o Polskę to nie jest paplanina na konferencjach prasowych. Ja PiS-u też nie kocham, ale kocham Polskę. Dlatego jako poseł niezależny apeluję do wszystkich posłanek i posłów, którzy kochają Polskę, aby okręt o nazwie Polska mógł przebić się przez rafy pandemii i rozwinąć żagle. Dziękuję, panie pośle. Proszę państwa, przystępujemy teraz do zadawania pytań. Pani marszałek.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Padają nieuzasadnione wątpliwości, że w razie bankructwa, inaczej niewypłacalności, jakiegoś kraju Unii Europejskiej reszta krajów członkowskich będzie obciążona spłatą zadłużenia tego kraju. Warto wspomnieć, że Unia Europejska w celu zapewnienia stabilności gospodarczej i finansowej stworzyła zbiór zasad ustanawiających nadzór gospodarczy i budżetowy dla całej Unii. Aby więcej nie było żadnych wątpliwości, proszę pana, panie premierze, o potwierdzenie, że Polska jest bezpieczna i nie będzie spłacać długów innych krajów. Dziękuję. Bardzo proszę panią poseł Izabelę Leszczynę, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Premier Morawiecki powiedział, że mamy dzisiaj podjąć ważną decyzję, i wyjątkowo nie skłamał.

Dlatego apeluję do PiS-u: odrzućcie swoje partyjne gierki, odrzućcie tak typową dla was chęć uwłaszczenia się na tych pieniądzach. Przyjmijcie poprawki Platformy Obywatelskiej. My nie chcemy wiele. Chcemy tylko, żeby obywatele mogli kontrolować, jak wydajecie te pieniądze, i żeby Sejm mógł kontrolować, czy realizujecie cele Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli przyjmiecie nasze poprawki, które nie są wygórowane, to zagłosujemy za Funduszem Odbudowy, ale jeśli chcecie uwłaszczyć się na tej kasie, tak jak robiliście to już wielokrotnie z wieloma funduszami, to nie będzie na to naszej zgody, bo to są pieniądze dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla samorządowców. I do dzisiaj ani samorządy, ani organizacje pozarządowe nie powiedziały wam: tak, nie dały wam zielonego światła.

Następne pytanie zadaje pani poseł Beata Maciejewska. Wysoka Izbo! Ta debata dzisiaj pokazuje, jak można patrzeć na interes Polski i Polaków. Tak robi np. Zbigniew Ziobro, który od lat wyklucza Polki i Polaków, który od lat np. ustami swoich przedstawicieli mówi, że polską racją stanu jest węgiel. który od lat wyklucza szeregi ludzi z polskiego społeczeństwa, który stoi, jest przeciwko ludziom.

Pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Panie Premierze! Pytanie moje kieruję do pana, panie premierze, w trosce o wiarygodność zobowiązań i obietnic, w tym również podanych na piśmie. Z jakim zdziwieniem czytałem krajowy program odbudowy, w którym okazało się, że po 5 latach jeździ ich ledwie 10 tys., 100 razy mniej niż obiecano.

Jak więc zatem my, parlamentarzyści i obywatele, którzy słuchają naszej debaty, mamy ufać i wierzyć panu w obietnicę wybudowania 75 tys. mieszkań? Może problemem jest również to, co zapisaliście w krajowym programie odbudowy: słaba jakość rządzenia. Pan poseł Artur Dziambor, koło Konfederacja. Panie Marszałku! Pan premier raczył tutaj sugerować, że Unia Europejska to taki Święty Mikołaj, który rozdaje prezenty, i one są bezpłatne, bezzwrotne. Faktycznie socjaliści tacy jak wy mogą jeszcze wierzyć w Świętego Mikołaja. Dojrzali politycy nie powinni być tak naiwni. Pan premier powiedział, że ten Fundusz Odbudowy to będzie szybki sposób na wyjście z kryzysu gospodarczego po COVID-19. A kto politycznymi decyzjami wprowadził nas w ten kryzys? Właśnie wy, właśnie wy. Dodrukowanymi pieniędzmi ratowaliście wybranych przedsiębiorców w tarczach antykryzysowych, a pożyczonymi pieniędzmi będziecie ratować spadające poparcie, oferując standardowo co? Łapówki ukryte pod płaszczykiem programów socjalnych. Niestety będzie trzeba to zgłosić w pewnym momencie do Trybunału Stanu.

Wysoka Izbo! 2050, Polska 2050, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Celem Funduszu Odbudowy jest nie tylko podniesienie gospodarki, ale także wspieranie tej gospodarki w kierunku przekształcenia w gospodarkę nisko-, bezemisyjną.

Przypomnę: co roku 50 tys. osób w Polsce umiera ze względu na jakość powietrza, płacimy jedne z najwyższych rachunków za prąd w całej Europie, a pan tego celu nie zadeklarował.

Mam krótkie pytanie do pana premiera: Czy zostały opracowane, czy zostaną opracowane jakiekolwiek obiektywne mierniki poprawy sytuacji, którą te środki mają nam przynieść?

Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Wielokrotnie w tej Izbie pan premier wspominał o rajach podatkowych, które ograbiają naszą gospodarkę. Mówił pan premier również o rajach podatkowych funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej, co jest wyjątkowym skandalem, pokazującym walkę poszczególnych państw o własne budżety, a nie o dobro Unii Europejskiej. Obecnie słyszymy jednak, iż Bruksela chce wycofać się z tego pomysłu, ulegając naciskom instytucji finansowych. Uprzejmie proszę o poinformowanie Polaków, czy, a jeżeli tak, to kiedy, ten podatek będzie wprowadzony. Dziękuję. Pani poseł Barbara Bartuś, klub Prawo i Sprawiedliwość. Nie, teraz nie pominąłem. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Nie, nie chce mi przejść, bo mi jest bardzo przykro, że państwo zajęliście się sobą i całkowicie zapomnieliście o Polakach i o potrzebach Polaków. Dlatego mam pytanie do pana premiera.

Dziękuję. Pan poseł Jacek Protas, Koalicja Obywatelska. Panie Premierze! Dużo pan ostatnio mówi o dobrej współpracy pana rządu z samorządowcami. Dlaczego zatem nie wsparliście naszej propozycji, ażeby z Krajowego Planu Odbudowy wydzielić pulę 40% środków i przeznaczyć ją na 16 koszyków regionalnych, którymi zarządzałyby samorządy województw? Przecież te samorządy udowodniły przez ostatnie lata, że potrafią transparentnie, zgodnie z zasadami i skutecznie zamieniać te pieniądze w pożyteczne dla społeczności lokalnych inwestycje. A wy postępujecie zupełnie odwrotnie. Chcecie pieniądze z grantów przeznaczyć dla spółek Skarbu Państwa, a samorządy nakarmić pieniędzmi z pożyczek. Samorządy muszą się zapożyczać na szpitale powiatowe, na inwestycje w kulturę, oświatę.

Panie Marszałku! Dziwi mnie, że sprawa ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy budzi takie kontrowersje i emocje. Dziwi mnie, bo rozmawiamy dzisiaj o gigantycznych środkach, które zadecydują o kondycji gospodarki polskiej w każdym aspekcie: lokalnym, krajowym, europejskim i światowym, i to nie na lata, ale na dekady. Dziwi mnie, że niektórzy chcą uzależnić wtłoczenie rzeki pieniędzy w europejski organizm gospodarczy, w każdy z jego krajów, od realizacji swoich osobistych, politycznych interesów. Ten fundusz będzie kształtował warunki życia Polek i Polaków, ale także wszystkich Europejczyków jeszcze wiele lat po tym, jak spory toczone dziś w tej Izbie ulecą w niepamięć. Pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję pani. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Panie Premierze! Apelował pan o solidarność w sprawie dochodów własnych Unii Europejskiej, tej decyzji, którą musimy tutaj zatwierdzić, ale oto podejmujemy tę decyzję w zupełnie przeciwny sposób. Najpierw mówimy o wydatkach, przesyłając Krajowy Plan Odbudowy do Brukseli bez konsultacji w Wysokiej Izbie, a dopiero później uchwalamy źródła finansowania.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska potrzebuje tych środków finansowych, to są ogromne fundusze, porównywalne z budżetem.

I będą zapewne dobrze zainwestowane, bo w systemie wydatkowania środków unijnych Polska zajmuje szóste miejsce na 27 państw. proszę pana ministra o informację, jakie mamy narzędzia zabezpieczające i gwarantujące, że te 770 mld zł zostanie przeznaczone na słuszne i właściwe cele. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.

Kto panu uwierzy? Kto uwierzy PiS, że będą dzielili pieniądze sprawiedliwie? To jest test na to, że państwo pokażecie: sprawiedliwie. Nikt. ...sprawiedliwie według PiS to fundusz inwestycji lokalnych - niektóre samorządy dostały pieniądze. Sprawiedliwie to 2 mld na telewizję publiczną, sprawiedliwie, a nie na ochronę zdrowia. A zatem, panie premierze, czemu państwo nie rozmawiali tu, na tej sali, czego państwo nie konsultowali w parlamencie? Jaki to był ciemny pokój, gdzie państwo zmusiliście Lewicę do tego, żeby się poddała? Państwo pokazujecie, że nie można wam wierzyć. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Chcę oświadczyć, że Lewicy nikt do niczego nie zmuszał. Chyba państwo widzicie, że jesteśmy tak samo traktowani jak wszyscy, czyli po minucie pan marszałek odcina nam mikrofon. Chcę zwrócić uwagę, szanowni państwo, na jedną rzecz. Otóż nigdzie w dokumentach Rady Europejskiej, w dokumentach Unii Europejskiej nie ma zapisu, że nieratyfikowanie tej umowy powoduje automatycznie odwołanie rządu jakiegokolwiek kraju. W związku z tym musimy Polkom i Polakom wytłumaczyć, że absolutnie ratyfikowanie tej umowy nie ma związku z upadkiem rządu. Po drugie, chciałbym się dowiedzieć od pana premiera, czy jest plan na najbliższy rok czy półtora roku, jeżeli chodzi o duże inwestycje, bo przecież prawie 50% tych środków jest przeznaczonych na ochronę klimatu, na elektromobilność. Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Drodzy Państwo! Rząd premiera Morawieckiego wykonał kawał dobrej roboty - wynegocjował 770 mld dla Polski. Wy tego nie chcecie. Nie chcecie tego? Nie chcecie? Nie chcecie tych pieniędzy? Nie chcecie na drogi, nie chcecie na cyfryzację, nie chcecie na innowacje? Nie chcecie tych pieniędzy. Proszę państwa, ja zagłosuję za.

i mieszkalnictwa w Krajowym Planie Odbudowy? Panie Premierze! Pan mówił dzisiaj w takim płomiennym proeuropejskim wystąpieniu, że pan jest za tymi pieniędzmi. Trzeba państwu wiedzieć, szczególnie państwu z Lewicy.

Panie Zandberg, ile mieszkań powstało za te 600 mld długu? Jak zmieniła się polska energetyka za te 600 mld? Pan powiedział tutaj dzisiaj w imieniu Lewicy, że to jest pchnięcie Polski w kierunku pogłębienia integracji europejskiej. Dzięki pana głosowi dzisiaj, w przyszłym tygodniu oni pchną integrację Polski z Unią Europejską, dzięki pani Pawłowicz, w drugą stronę. Pan powiedział, że to jest pociąg do Europy. Pan pociąg z kibitką pomylił. Pan poseł Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiemy dobrze, iż Krajowy Plan Odbudowy był bardzo szeroko konsultowany. Chciałbym zapytać, panie premierze, kto brał udział, kto wziął udział w tych konsultacjach i jaki był wynik tych konsultacji. Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W debacie nad Funduszem Odbudowy i Krajowym Planem Odbudowy kompletnie zapomnieliśmy o tym, że jako Europejki i Europejczycy stworzyliśmy plan odbudowy po pandemii jako most od kryzysu do zielonej i innowacyjnej gospodarki, a przysłany wczoraj do komisji dokument nie jest takim mostem. On nie jest nawet chybotliwą kładką. Wiele inwestycji wpisanych w KPO jest niezgodnych z zasadą: nie czyń poważnej szkody, i może doprowadzić do degradacji środowiska. To nie jest Krajowy Plan Odbudowy, to jest krajowy plan zmarnowanej szansy. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W przestrzeni publicznej pojawiają się często informacje, że oto będziemy mieli do czynienia z uwspólnotowieniem zobowiązań w sytuacji, gdyby któreś z państw członkowskich nie spłaciło pożyczki gwarantowanej przez Unię Europejską. Dlatego mam pytanie, panie premierze. Czy prawdą jest, że decyzja, którą mamy ratyfikować, ustala górny pułap wpłat do budżetu Unii Europejskiej dla każdego państwa niezmiennie wobec jakichkolwiek okoliczności w przyszłości? Czy prawdą jest, że jest to uregulowane nie tylko w pakiecie budżetowym, ale ma też odzwierciedlenie w akcie wyższego rzędu, to jest w art. 125 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie wprost jest powiedziane, że nie jest możliwe przejęcie zobowiązań jednego kraju przez drugi? Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Nie zagłosuję przeciw, bo uważam, że Fundusz Odbudowy jest jedyną szansą na ożywienie europejskiej gospodarki i Polska oczywiście musi brać w tym udział. Ale nie będę za, dlatego że pański rząd nie zrobił nic, aby wyjaśnić jakąkolwiek aferę, gigantyczne przekręty na gigantyczne pieniądze - i żadnego winnego.

i ostatniej afery - wyborów kopertowych. Publiczne pieniądze są od jakiegoś czasu poza jakąkolwiek kontrolą.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Polska racja stanu wymaga tego, aby polski Sejm ponad podziałami ratyfikował umowę o Funduszu Odbudowy. Panie Premierze! Dziękując panu za dobre brukselskie negocjacje, za duże pieniądze, które wynegocjował pan dla Polski, chciałem zapytać: Czy uzasadniona jest teza głoszona przez część opozycji, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy spowoduje ustanowienie nowych podatków krajowych w Polsce? Czy ta teza jest prawdziwa czy to jest po prostu zwykła manipulacja totalnej opozycji, która jest wrogo nastawiona do rządu Prawa i Sprawiedliwości? Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Ale mam dla pana złą wiadomość. Niestety nie uda się panu uzyskać tych 770 mld, którymi się pan chwali, a zwłaszcza 250 mld z Krajowego Planu Odbudowy, po prostu dlatego że propozycje zgłoszone do Brukseli nie spełniają wymaganych kryteriów. Jednym z tych kryteriów jest zalecenie ze strony Komisji Europejskiej i Rady z maja ubiegłego roku o tym, żeby poprawić klimat inwestycyjny, a środkiem do tego ma być wzmacnianie niezależności sądów. Chcę więc panu powiedzieć, że na 500 stronach tego dokumentu, który wysłaliście do Brukseli, ani razu nie pojawia się pojęcie niezależności sądów. Pani poseł Teresa Wargocka, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata nad środkami unijnymi dla Polski jest bardzo burzliwa.

Wszystkie zarzuty o to, że środki mogą być zmarnowane, zdefraudowane, wykorzystane politycznie, są naprawdę obraźliwe.

Te środki zawsze były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pani poseł Maria Janyska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, pani poseł.

Wysoka Izbo! Pan premier, grając na emocjach, dzisiaj kilkakrotnie przywoływał polską rację stanu. A jak wygląda polska racja stanu w waszym wykonaniu? Kilka obrazów z dzisiaj.

Przedstawiciel pracodawców informuje, że Rada Dialogu Społecznego nie otrzymała ostatecznej wersji KPO, a to Rada Dialogu Społecznego opiniuje projekty rządowe. Znów pominięcie. KPO jak nie zawierał, tak nie zawiera kryteriów zasad jawności, przejrzystości i sprawiedliwości rozdawania pieniędzy. Ale my was uratujemy. Pan poseł Sylwester Tułajew, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Historyczna chwila, przed którą stoi Polska. Historyczna chwila, przed którą stoi polski parlament. Dziś zdecydujemy, czy skutecznie i sprawnie wrócimy na drogę, na ścieżkę rozwoju, czy też w imię kompletnie niezrozumiałych zagrywek partyjnych Koalicji Obywatelskiej nie skorzystamy z tej szansy. Chciałbym zaapelować do posłów Platformy Obywatelskiej, a w sposób szczególny do posłów Platformy Obywatelskiej z województwa lubelskiego, aby zagłosowali za tą ustawą, aby zagłosowali za 40 mld zł dla naszego regionu. Dzisiaj warto również zapytać, by po raz kolejny wyjaśnić bardzo prostą sprawę, czy od ratyfikacji zależy całość finansowania z Funduszu Odbudowy i czy ta ratyfikacja jest związana z całym funduszem unijnym. Dziękuję bardzo.

Kilka lat temu z tego miejsca pan premier Morawiecki przedstawiał swój plan, plan Morawieckiego, „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Nic z tego planu nie zrealizował. Zostały tylko slajdy. Dlaczego nie zrobił niczego? Bo po prostu rozkradliście Polskę. Ale panu nie wolno wierzyć, bo

Panie premierze, to nie jest żaden plan Marshalla.

Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Podczas dyskusji nad strukturą wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy pojawiły się wątpliwości co do wysokości środków finansowych adresowanych do rolników i przemysłu rolno-spożywczego. Z tych środków ma być finansowany komponent pod nazwą: inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inwestycje w tym programie obejmą szerokie spektrum sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowane formy współpracy rolników, spółdzielnie oraz podmioty gospodarcze z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Pan poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako długoletni samorządowiec, będąc parlamentarzystą, nadal bardzo blisko współpracuję z koleżankami i kolegami samorządowcami, i to z różnych opcji, co chcę podkreślić i mocno zaznaczyć. Pamiętam też, że nie było tak szerokich konsultacji przy poprzednim budżecie unijnym. Nasz wpływ był w zasadzie bliski zeru. W związku z powyższym mam pytania: Czy będzie, a jeżeli tak, to jak będzie wyglądała, dalsza praca komisji wspólnej rządu i samorządu? Czy prawdą jest, jak twierdzi, chciałoby się powiedzieć, totalna opozycja, ale przepraszam, fakt jest taki, że coraz mniej znacząca, mała opozycja, że samorządy nie będą miały już nic do powiedzenia? Pytam się: Czy samorządy będą współdecydowały, będą partnerem dla rządu?

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Dziś mamy bardzo ważny dzień dla Polski, można śmiało powiedzieć, że historyczny dzień dla Polski, ponieważ w polskim parlamencie możemy uruchomić 770 mld zł dla Polski, dla naszej ojczyzny. Ten dzień i to głosowanie będą również szczególnie ważne, jeśli chodzi o pokazanie wiarygodności i braku wiarygodności każdego polskiego parlamentarzysty. Pamiętajcie, szanowni państwo, panie i panowie posłowie z Platformy Obywatelskiej, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.

Pan poseł Zdzisław Sipiera, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! O tym, że wydajemy środki na duże inwestycje, wszyscy wiemy. To gołym okiem jest widoczne, kiedy przez Polskę przejeżdżamy. Ale są też bardzo istotne inwestycje regionalne. Takich środków, jakie w ostatnich latach otrzymują samorządy, nigdy nie było. To jest fakt, który ma miejsce tu i teraz.

I moje pytanie jest właśnie takie: Jak to będzie się odbywało w najbliższym czasie? Czy te inwestycje w koleje regionalne będą w najbliższym czasie się odbywały? Pan poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoki Sejmie! Krajowy Plan Odbudowy to przełomowy moment w historii Polski, to realna szansa wzmocnienia Polski pokoleniowej, silnej, bezpiecznej i nowoczesnej. Jednym z głównych filarów jest ochrona zdrowia, zatem zwiększenie kadry medycznej, zwiększenie naboru na studia medyczne. To nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa.

To telemedycyna. To prawie 30 mld zł, łącznie z europejskim instrumentem na rzecz spójności terytorialnej. Zatem kto nie zagłosuje za środkami unijnymi i za Krajowym Planem Odbudowy, jest przeciw Polsce, jest przeciw zjednoczonej Europie. Tym razem Polak musi być mądry przed szkodą.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Celem polityki jest realizacja dobra wspólnego wszystkich obywateli. To dzisiejsze głosowanie jest szansą rozwojową Polski na lata. Taka sytuacja w tej Izbie powinna nas wszystkich łączyć. Od paru dni Platforma Obywatelska próbuje utrudnić przyjęcie tych środków. Dziś od rana są wnioski o przerwę, wnioski o odroczenie obrad. Platforma Obywatelska dziś mówi Polakom wprost, że w najbliższych latach ma być bieda, bo tylko w taki sposób widzicie swoją szansę na dojście do władzy. To niespotykana sytuacja w polskiej polityce. PiS, będąc w opozycji, zawsze wspierało rząd, bo taka jest racja stanu. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Szanowni Państwo!

Skutki pandemii, już wtedy widoczne, były na tyle poważne, że należało szukać ekstraordynaryjnych rozwiązań. Zaraz po tym przystąpiliśmy do prac nad Krajowym Planem Odbudowy.

Od pierwszego dnia był zaproszony, dokładnie tak samo jak premier, wicepremierzy, ministrowie rządu, którzy uczestniczyli w prezentacji Krajowego Planu Odbudowy. Już wówczas była możliwość dyskutowania o Krajowym Planie Odbudowy. Co się wydarzyło od tamtego czasu? Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań, w których uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora, przedsiębiorcy. Wszyscy zainteresowani mogli zabrać głos. Polacy, zwykli Polacy pisali do nas z uwagami. Myśmy wszystkie przeczytali. Staraliśmy się je przeanalizować, wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy. Kilkaset uwag realnie udało się wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy. Jest to 30 kwietnia.

I co się, szanowni państwo, okazuje? Po tym czasie, dopiero 4 maja, największa partia opozycyjna mówi, że ma propozycje i poprawki, i jest oburzona tym, że nie możemy ich nanieść na Krajowy Plan Odbudowy. byliśmy gotowi i chętni dyskutować o państwa poprawkach, tylko ich po prostu nie było. W marcu Lewica, ale również koło 2050 złożyły na piśmie poprawki. Był przedmiot do negocjowania, do spotykania się. Państwo takiej szansy sobie nie daliście. Szanowni Państwo! Słuchałem każdego z wystąpień i powiem państwu szczerze: nie wiem, dlaczego państwo są przeciwni. Nie padł żaden argument, który by wskazywał merytoryczne uzasadnienie wniosku o wstrzymanie się albo bycie przeciwnym. Były głosy za, były głosy, które wskazywały na jakieś uwagi ze strony Konfederacji. Państwo wykazali jedno: są przeciwni Prawu i Sprawiedliwości i tylko dlatego zagłosują przeciwko. Tylko dlatego. Odnosząc się do uwag, powiem państwu szczerze, że tak już zupełnie po ludzku przykro mi jest słuchać tego, jak państwo się odnoszą do przedstawicieli Lewicy. Mówił o przyjacielach 276. Mówił o grupie, która przejmie władzę. Nie minęły 2 miesiące i państwo ich obrażają na każdym kroku. To są partnerzy do rozmów? Odpowiadając na pytania, które pojawiły się w trakcie dyskusji.

Uczestnictwo samorządów w realizacji środków europejskich.

Tutaj w najmniejszym stopniu tego nie zmieniamy. Oczywiście beneficjentami środków również będą samorządy. Na dzisiaj informacja jest taka, że ostateczny plan przewiduje grubo ponad 30% na rzecz samorządów. Zaczynaliśmy od poziomu 17%, ale uwagi, konsultacje, rozmowy z samorządowcami doprowadziły do sytuacji, w której dziś mamy trzydzieści kilka. I mogą państwo dzisiaj powoływać się na samorządowców, ale to myśmy z nimi rozmawiali i myśmy słyszeli, co oni mówili: my popieramy Krajowy Plan Odbudowy, tylko boimy się to publicznie oświadczać. Bo państwo na nich nacisk stosują. Państwo mówią: bądźcie przeciwko, bo nie będziecie z nami. Nawet prezydenci dużych miast spotykali się z nami. Przyjeżdżali i pytali o konkretne inwestycje. Pytali o metro, pytali o tramwaje. Były takie uwagi. Ostatni raz pana ostrzegam, panie pośle.

Oczywiście tę regułę spełniamy. Zamówiliśmy niezależną analizę, która ocenia wszystkie projekty, które są ujęte w Krajowym Planie Odbudowy, i mamy analizę, którą przesłaliśmy łącznie z ostatecznym planem odbudowy. Tereny wiejskie i rolnictwo, szanowni państwo, samorządy i rolnictwo to są dwa obszary, które najwięcej zyskały w wyniku konsultacji. Byli najbardziej aktywni i największe przesunięcia zrobiliśmy na ich rzecz.

Takich środków ponad WPR i ponad PROW na polskiej wsi nie było.

Ale też muszę uczciwie powiedzieć, że rozmawialiśmy na temat wielu spraw z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiele uwag również tutaj uwzględnialiśmy. Szanowni Państwo! Za 10 lat prawdopodobnie większości z nas tutaj, w parlamencie, nie będzie. Ale będzie informacja o tym, jak który poseł zachował się przy tej bardzo ważnej decyzji IX kadencji. Nie dajcie sobie wmówić, że Borys Budka decyduje, jak macie głosować.

które wychodzą naprzeciw polskim potrzebom rozwojowym w tym szczególnym czasie - w szczególnym czasie, w którym znalazła się Unia Europejska. Ja chciałbym się odnieść do tych uwag - wypowiadanych czasem w bardzo dramatycznym tonie, choć nie zawsze poważnym - które odnoszą się do kwestii suwerenności, do kwestii europejskiego opodatkowania, w końcu do kwestii uwspólnotowienia długu. Powiem szczerze, że gdyby te oceny, które padły na tej sali z ust prawicowej opozycji, miały cokolwiek wspólnego z prawdą, to sam bym protestował, ponieważ nie jestem zwolennikiem Europy federalnej, ponieważ nie uważam, aby dla Europy dobrym rozwiązaniem było uwspólnotowienie długu, ponieważ nie uważam, aby rozwijanie kompetencji fiskalnych Unii Europejskiej było właściwą odpowiedzią na problemy, które mamy przed sobą. Ale tak nie jest. Dlatego z czystym sumieniem mogę państwa zachęcać kolejny raz do tego, aby tę misterną konstrukcję, tę bezpieczną dla polskich finansów publicznych konstrukcję poprzeć. Zagwarantowaliśmy nie tylko olbrzymi zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki, który wyjdzie naprzeciw tym wszystkim potrzebom, które już dziś są palące, a za rok mogą być jeszcze bardziej palące. Premier Morawiecki zagwarantował nie tylko zastrzyk pieniędzy, ale również gwarancje prawno-instytucjonalne dla bezpieczeństwa finansów publicznych Polski. Powiem państwu, że Polska nie jest w tej sprawie osamotniona. Jest bardzo niewiele państw, na palcach jednej ręki można zliczyć państwa, które na serio życzyłyby sobie uwspólnotowienia długu. Znakomita większość państw, podobnie jak Polska, nie życzy sobie uwspólnotowienia długu. Dlatego takie ryzyko jest całkowicie abstrakcyjne. Takiego ryzyka po prostu nie ma. Zadbaliśmy również o to - chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno, ponieważ ta sprawa powraca jak bumerang - aby odrzucić opodatkowanie europejskie oparte o przychody z systemu emisji

Tak długo, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie zgody na podatki europejskie o regresywnym charakterze. Wbrew temu, co padało na tej sali - po wielu przecież miesiącach, kiedy można było przestudiować wyniki negocjacji, konkretne projekty decyzji, także tę decyzję, której ratyfikacją mamy się zająć właśnie teraz - nie ma decyzji w sprawie podatku od transakcji finansowych, nie ma decyzji o podatku dotyczącym gospodarki cyfrowej. Nie ma, aczkolwiek Polska pozostaje aktywnym, konstruktywnym uczestnikiem tej debaty, ponieważ niektóre formy tego podatku mogłyby spowodować, że ciężar finansowania Unii Europejskiej byłby lżejszy dla Polski, a cięższy dla innych gospodarek. Wydaje się, że nie ma sensu prowadzić doktrynalnej tępej dyskusji na temat tego, czy to dobrze czy źle, tylko jest sens skupić się na tym, czy to się opłaca, czy to też się nie opłaca. W tej dyskusji Polska uczestniczy bardzo aktywnie od wielu lat. To nie tylko kwestia przywołanego tutaj traktatu, który wyraźnie, czarno na białym jako ustawa zasadnicza Unii Europejskiej zabrania przenoszenia odpowiedzialności za czyjekolwiek długi. Możecie państwo to przeczytać w samej decyzji, o której tutaj dzisiaj mowa, możecie państwo o tym przeczytać w konkluzjach z lipca i grudnia, możecie w końcu państwo o tym przeczytać w bardzo obszernej oficjalnej analizie służb prawnych Rady Unii Europejskiej.

Skoro państwo są tym tak zainteresowani, to myślę, że warto byłoby rzucić okiem na dokumenty, w szczególności na opinie służb prawnych Rady, ponieważ tam to jest napisane czarno na białym, nie tylko pod kątem naszych potrzeb, naszych oczekiwań, tego, w jaki sposób my rozumiemy te decyzje, ale również pod kątem interesów i oczekiwań całej długiej listy państw, znakomitej większości państw, które tak jak Polska nie życzą sobie uwspólnotowienia długu Unii Europejskiej.

Ale nawet gdyby się okazało, że któreś z państw członkowskich bankrutuje, wycofuje się z rynku, przestaje płacić zobowiązania, to nadal zobowiązania związane z tą decyzją pozostają zobowiązaniami tego państwa. I nikt - ani Unia, ani inne państwo członkowskie - takiego zobowiązania przejąć nie może. Nie jest to kwestia decyzji politycznej, tylko kwestia ograniczeń natury prawnej. Krótko mówiąc, pamiętajmy o jednej rzeczy: ta decyzja i ta debata nie dotyczy tylko tego, że Polska ma szansę na to, żeby efektywnie sięgnąć po bardzo duże środki na swoje bardzo konkretne potrzeby rozwojowe tu i teraz, ona również stanowi wręcz gwarancję bezpieczeństwa fiskalnego Polski na przyszłość.

Jest ona bezpieczna dla Polski pod każdym względem. Ostatnia sprawa. Najbogatsze państwa członkowskie Unii Europejskiej od lat szukają dobrego pretekstu, dobrego wytłumaczenia, jak by tu mniej płacić na Unię Europejską. W jakimś sensie jest to zrozumiałe, aczkolwiek myślę, że bardzo krótkowzroczne, ponieważ przez to Unia się nie rozwinie, Unia nie będzie mogła odpowiadać na realne potrzeby Europejczyków. Są to państwa, które często się powołują na swój nieprawdopodobnie proeuropejski etos, a jednocześnie chcą płacić mniej na Unię Europejską. Szukają wymówki. Jedną z takich wymówek jest oczywiście monetaryzm, państwo minimum, czasami, jak w przypadku niektórych niemieckich ośrodków, zasada demokratycznej kontroli Bundestagu nad budżetem, nad zobowiązaniami państw.

To są działania, które są wprost wymierzone w interesy rozwojowe Polski.

Wszystkie korzyści ze wspólnego rynku, także płynące z polskiej rozwijającej się gospodarki, bierzemy, nie płacimy na budżet europejski po to, aby model rozwoju zależnego był utrzymywany tak długo, jak się da. Aby państwa Europy Środkowej nie emancypowały się gospodarczo, aby nie rozwijały się gospodarczo w taki sposób. aby być podmiotem, prawdziwym podmiotem. Tu dochodzimy do kwestii zasadniczej. Jakie są wymiary suwerenności? Czy suwerenności przybywa od tego, że o niej mówimy, że o niej krzyczymy? Czy też suwerenności przybywa, także Polsce, od tego, że jesteśmy silniejszą gospodarką, silniejszym państwem, że się rozwijamy.

W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania po doręczeniu posłom zestawienia zgłoszonych poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Ogłaszam przerwę do godz. 19.15.

który kilkakrotnie okłamał Wysoką Izbę. Chciałabym przypomnieć panu ministrowi, że miejscem na debatę pomiędzy opozycją a stroną rządząca jest Sejm: sala plenarna i posiedzenia komisji. Chciałabym przypomnieć, że klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o informację bieżącą. Nasi posłowie złożyli pięć wniosków o zwołanie pięciu posiedzeń komisji, [[Oklaski]] na których składaliśmy wnioski, na których mówiliśmy, co jest w tym Krajowym Planie Odbudowy złego. Dlatego chcę wyraźnie powiedzieć, że klub Koalicji Obywatelskiej jako jedyny w pierwszym czytaniu złożył sześć poprawek, które gwarantują kontrolę społeczną nad wydawaniem pieniędzy, kontrolę Sejmu nad realizacją celów KPO.

Proszę państwa, ponieważ za chwileczkę będziemy głosować, to teraz przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa obecnych na sali i tych, którzy są z nami połączeni zdalnie, o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na głosowaniach. Bardzo proszę.

Oczywiście, proszę państwa, wznowiłam obrady.

Stwierdzam kworum. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1131) Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1131, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Wobec propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu zestawienia poprawek zgłoszono sprzeciw, który rozstrzygniemy w głosowaniu. Odrzucenie tej propozycji będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu zestawienia poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm propozycję przyjął. W trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono poprawki. Sejm podjął decyzję o nieodsyłaniu projektu ustawy do komisji i o przystąpieniu do głosowania po doręczeniu paniom i panom posłom tekstu poprawek. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1123. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie zgłoszone w drugim czytaniu poprawki. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują, aby dodać preambułę do ustawy.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił. W 3. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują m.in., aby Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności przyjmowany był w drodze ustawy.

W 4. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują m.in., aby w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności wyodrębnić 16 koszyków regionalnych. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

W 5. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują m.in., aby określić zasady wyboru projektów do dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

W 6. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują, aby utworzyć Komitet Sterujący nadzorujący realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz określić m.in. jego skład i kompetencje. Głosujemy.

W 7. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują m.in., aby określić odrębne zasady uczestnictwa w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności podmiotów, o których mowa w tym przepisie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

W 8. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują, aby po ratyfikacji przedmiotowej decyzji Rady zobowiązać Radę Ministrów do podjęcia działań w celu notyfikowania zamiaru przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 9. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują, aby Sejm zobowiązał Radę Ministrów do przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej.

Tak że spokojnie.

W 10. poprawce wnioskodawcy w dodawanym artykule proponują, aby Sejm zobowiązał Najwyższą Izbę Kontroli do corocznej analizy wydatkowania środków, o których mowa w tej propozycji.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1123, zechce nacisnąć przycisk.

Proszę usiąść na miejsce. Nie, przykro mi bardzo, ale jesteśmy w trakcie głosowania.

Pan jest konstytucjonalistą? Nie wiedziałam, panie pośle.

To ma jeszcze szansę. Proszę państwa, jak się korzysta z tabletu, prowadząc, to nie jest to takie proste, bo on mi się ciągle wyłącza. Ale państwo macie tylko do pstrykania, a ja mam do prowadzenia i do stukania.

Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo!

Dopuszczone zostały do głosowania, co nie zmienia faktu, że z dwóch powodów poprawki do ustawy ratyfikacyjnej nie są przyjmowane. Po pierwsze, dlatego że. nie dopuszcza tego polska procedura legislacyjna. Po drugie, zwracam uwagę, że w tych 19 krajach, które do tej pory ratyfikowały, żadna ustawa ratyfikująca tę decyzję nie jest opatrzona warunkami. Dziękuję bardzo.

Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Taki, że to jest minister, któremu udzieliłam głosu. Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą.

Oświadczenie? Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Odnośnie do wystąpienia pana ministra Wawrzyka: Sejm jest gospodarzem ustaw. Sejm jest. Często używane przez was słowo „suweren” trzeba przypomnieć. Jest on wybrany przez suwerena i ma prawo decydować o kształcie każdej ustawy. Preambuła jest naszą intencją, jest wyrażeniem woli, jest pokazaniem kierunku, w którym Fundusz Odbudowy ma zmierzać. Nie zdecydowaliście się go poprzeć, nie wiem, z obawy przed tym, że. Nie wymigujcie się teraz, bo ograniczacie tym samym suwerenność Sejmu Rzeczypospolitej: w przyjmowaniu ustawy, w przyjmowaniu najważniejszych aktów. Przyjmiemy tę preambułę w Senacie. Pani poseł Agnieszka Soin, klub Prawo i Sprawiedliwość, z oświadczeniem. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, który przypada dzisiaj, pragnę podziękować wszystkim pełniącym tę zaszczytną i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszom, zarówno z państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej, za ich zaangażowanie i wkład pracy. Dziękuję też ich rodzinom za udzielenie im emocjonalnego wsparcia oraz za przyzwolenie na codzienne poświęcenie, a często też narażanie życia. Chciałabym przy tej okazji wyszczególnić Ochotniczą Straż Pożarną w Twardogórze w województwie dolnośląskim, gdzie sprawuję mandat poselski, Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze istnieje od 1945 r., gdy na wniosek burmistrza 29 października wybrano jej władze. Od 75 lat miasto Twardogóra, ja i sąsiadujące z nią miejscowości mogą liczyć na pomoc strażaków w miejscowych zagrożeniach, alarmach oraz pożarach. Dziękuję obecnemu zarządowi oraz członkom remizy, którzy kontynuują tak ważną dla nas służbę i kultywują strażacką tradycję niesienia pomocy: panu prezesowi Tomaszowi Dżugajowi, jego zastępcy Ireneuszowi Mimietzowi, naczelnikowi Marcinowi Badowskiemu, jego zastępcy Krzysztofowi Szostkowi, skarbnikowi Małgorzacie Olszańskiej, sekretarzowi Marcinowi Kiełtyce, gospodarzowi Tomaszowi Małaniakowi oraz członkom Krzysztofowi Małaniakowi i Grzegorzowi Blaźniakowi. Dziękuję bardzo, pani poseł. Kolejne oświadczenie, pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Zapraszam, panie pośle. Szanowny Panie Premierze! Zaszczep się w majówkę, w mobilnych punktach ustawionych w 16 stolicach polskich województw. W województwie kujawsko-pomorskim, w którym od ponad 20 lat są dwie równorzędne stolice, w Bydgoszczy i Toruniu, zorganizowano jeden punkt szczepień w Toruniu. W związku z powyższym mieszkańcy Bydgoszczy za moim pośrednictwem kolejny raz pytają: Co politykom Prawa i Sprawiedliwości zrobiła Bydgoszcz, że nawet w organizacji akcji szczepień funkcjonariusze rządu bez cienia żenady pokazują, że dla rządu jesteśmy miastem drugiej kategorii? Być może jacyś politycy w Warszawie cieszą się z tego, że przy ich szczepieniach jesteśmy.

Szanowny Panie Premierze! Od wielu miesięcy województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z pierwszych miejsc w Polsce w statystykach umieralności na COVID, o czym przypomniałem ministrowi zdrowia w mojej interpelacji poselskiej. Dlatego było pełne uzasadnienie epidemiczne, by mobilne punkty szczepień stanęły i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a nawet w mniejszych miejscowościach naszego regionu. Do wsparcia takiej akcji w Bydgoszczy był gotowy duży powszechny punkt szczepień w centrum targowym w Myślęcinku. Są województwa, w których rząd właśnie tak zorganizował majowe szczepienia w kilku punktach. Dla mieszkańców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego tej życzliwości i pozytywnych działań ze strony rządu niestety zabrakło. W związku z opisanymi faktami chciałem zwrócić się i zwracam się do pana premiera z prośbą o udzielenie pilnej odpowiedzi na piśmie na pytanie: W jaki sposób i kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zorganizuje dodatkową akcję szczepień w Bydgoszczy dla mieszkańców miasta oraz dla miast i gmin bydgoskiego obszaru funkcjonalnego, niezależnie od zaplanowanych i zrealizowanych na dzień dzisiejszy szczepień systemowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj szczególny dzień. 4 maja wspominamy i świętujemy to wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień strażaków. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim druhom strażakom z ochotniczych straży pożarnych. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej za olbrzymie zaangażowanie. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że każdego dnia strzegą bezpieczeństwa Polaków, strzegą bezpieczeństwa obywateli.

Trzeba przypomnieć wielki program modernizacji służb mundurowych. To właśnie z tego programu na państwową straż pożarną wydatkowaliśmy w ostatnich latach 1700 mln zł, z czego prawie 500 mln zł zostało przeznaczone na ochotnicze straże pożarne. Dziękuję za to, że bardzo często jesteście pierwsi wtedy, kiedy ludzie potrzebują waszej pomocy, a szczególnie w tym ostatnim czasie, czasie pandemii. Za to, drodzy strażacy, wam bardzo serdecznie dziękuję.

Funkcjonariusz Policji, który na służbie wykonywał swoją powinność, podejmował interwencję, został postrzelony przez bandytę. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych bohaterach w mundurze, chciałbym, żebyśmy oddali cześć temu wyjątkowemu funkcjonariuszowi, który do końca zrealizował ślubowanie policyjne, który zginął na służbie. Chciałbym przekazać kondolencje wszystkim funkcjonariuszom, ale przede wszystkim rodzinie. I chciałbym zapewnić, że jako parlamentarzyści. Ale również wiem o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmie się rodziną, zaopiekuje się nią w sposób odpowiedni. I proszę Wysoką Izbę, abyśmy uczcili chwilą ciszy zmarłego dzisiaj policjanta, który został zabity przez bandytę w Raciborzu. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Bardzo proszę.

Panie Premierze! Panie Ministrze Rolnictwa! Wysoka Izbo! Dziś branża drobiarska przeżywa bardzo głęboki kryzys.

W kraju wykryto do tej pory 265 ognisk ptasiej grypy. Rok wcześniej było ich zaledwie 35. Do dzisiaj zutylizowano 10 mln sztuk drobiu: 5 mln sztuk kur niosek, 1,1 mln brojlerów, ponad 1 mln indyków, zlikwidowano pojedyncze stada gęsi i kaczek. W budżecie na rok 2021 na zwalczanie chorób zakaźnych przewidziano 430 mln zł. Do tej pory straty wyliczone tylko w powiatach żuromińskim, mławskim i sierpeckim wojewódzki lekarz weterynarii wycenił na 500 mln zł. Szanowni Państwo! Panie Premierze! Potrzebna jest pilna nowelizacja ustawy, bo nie policzyliśmy tutaj Warmii i Mazur, nie policzyliśmy Wielkopolski, nie policzyliśmy Kujaw, nie policzyliśmy reszty kraju. Te straty znacznie przekraczają 430 mln zł. Rolnicy borykają się z ogromnymi problemami, mają potężne problemy, zatory płatnicze. Po pierwsze, nie mogą zapłacić za pisklęta, za paszę, za prąd. Nie posiadają pieniędzy na obsługę kredytów bankowych. Kolejnym ciosem jest utylizacja jaj, paszy i obornika. Rolnicy, którzy mają zdrowe stada, nie wiedzą, czy kupować paszę czy hodować dalej, czy w ogóle ich ptaki będą utylizowane. Dzisiaj w powiecie Ostrów Wielkopolski przeznaczono do utylizacji kolejne 150 tys. sztuk. Potrzebne jest pilne zwołanie komisji rolnictwa, poznanie właściwych strat podanych przez lekarzy wojewódzkich i powiadomienie rolników, kiedy otrzymają należne im odszkodowania. Należy też pamiętać o lekarzach weterynarii, którzy zostali skierowani do pracy z różnych rejonów kraju. Dzisiaj pan minister Waldemar Buda prosił posłów PSL o właściwe głosowanie: za Funduszem Odbudowy.

Bardzo proszę. Panie Przewodniczący Komitetu Kaczyński! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak to jest, że pieniądze z Funduszu Odbudowy prawie dla wszystkich europejskich krajów oznaczają święto radości, nadzieję na powrót do normalności po tak trudnym pandemicznym czasie? Powinnam się dziś cieszyć, z wielką radością iść do Sejmu i jako Europejka bez chwili zawahania zagłosować za uruchomieniem tych środków. A jednak przez partię rządzącą nie mogłam tego zrobić. Bo nie spojrzałabym sobie w oczy, gdybym miała na sumieniu miliardy złotych, które nie trafią do wszystkich Polek i Polaków, a staną się funduszem wyborczym PiS. Tylko u nas rządzący nie chcą sprawiedliwie rozdać tych pieniędzy, tak by trafiły do wszystkich obywatelek i obywateli. Wręcz przeciwnie, robią wszystko, by oszukać Unię, a środki zawłaszczyć, np. przez ogromne dotacje bezzwrotne dla spółek Skarbu Państwa - przypomnę, że samo PGE złożyło wnioski na 74 mld zł, czyli 35% całego funduszu - rozdać swoim, jak w przypadku pieniędzy z funduszów lokalnych, które trafiły tylko do PiS-owskich samorządów, źle ulokować, jak już to bywało z bezużytecznymi maseczkami, albo zgubić, jak dzisiaj 700 tys. szczepionek. Kto bogatemu zabroni? Doprowadziliście do tego, że głosowanie nad nimi stało się jątrzącą raną i nie ma właściwie z tej sytuacji dobrego wyjścia. Zagłosowaliście za? To daliście przyzwolenie na fundusz wyborczy dla PiS-u, na olbrzymie dotacje dla państwowych spółek Skarbu Państwa, na dalsze zadłużanie samorządów, bo będą one mogły korzystać tylko z części pożyczkowej. Wstrzymaliśmy się? To jedna strona oskarży nas o zbyt mało wyraziste zdanie, a druga i tak będzie wypominać, że nie było poparcia. A może zagłosowaliście przeciw? To będzie zarzut, że jak możecie zabierać tę kasę ludziom. Wybór dosłownie jak w greckiej tragedii. Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oświadczenie w sprawie sprawiedliwego handlu. Sprawiedliwy handel to oddolny międzynarodowy ruch społeczny, którego celem jest poprawa warunków życia drobnych producentów kawy, herbaty, kakao, cukru, bananów i innych produktów z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej mogą godnie pracować, otrzymywać uczciwą cenę za wytwarzane produkty, ale mogą też nawiązywać sprawiedliwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch sprawiedliwego handlu tworzony jest przez organizacje pozarządowe, wolontariuszy, działaczy oraz firmy przy udziale świadomych konsumentów. Wdrażanie zasad sprawiedliwego handlu ma realny wpływ na rozwiązywanie problemów ubóstwa, pracy niewolniczej, wykorzystywania do ciężkiej pracy dzieci, braku dostępu do rynków zbytu oraz uzależnienia od pomocy otrzymywanej z tzw. krajów wysoko rozwiniętych. W XXI w. sprawiedliwy handel winien stać się najbardziej rozpoznawalną formą pomocy rozwojowej dla krajów ubogiego południa. Sprawiedliwy handel to nie tylko wymiana handlowa, ale znacznie szersza idea sprawiedliwości w handlu światowym. Produkty sprawiedliwego handlu oznaczone są międzynarodowym znakiem systemu certyfikacji fair trade. Oferta tych produktów oraz sieć ich dystrybucji dzięki coraz większej świadomości konsumentów stale się powiększają. W Polsce jest zaledwie kilka miast, które mogą pochwalić się tym zaszczytnym tytułem. Z prawdziwą dumą mogę powiedzieć, że wśród nich jest moje miasto, Jelenia Góra, które jako drugie w Polsce uzyskało ten tytuł w 2018 r.

Apeluję, zachęcam panie i panów posłów oraz władze samorządowe wszystkich szczebli do zaangażowania się w wielką ideę międzynarodowej solidarności z mieszkańcami ubogich krajów w ramach ruchu sprawiedliwego handlu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Ostatnie dni kolejny raz utwierdzają Polki i Polaków w przekonaniu, że czegokolwiek dotknie się PiS-owski rząd, to to spartaczy. Przypomnę, że przed długim majowym weekendem minister Michał Dworczyk ogłosił, że czeka nas wielka majówka pod hasłem: Szczepmy się. Powiem państwu, jak ona wyglądała w Lublinie, moim rodzinnym mieście. Otóż na jednym z głównych placów miasta, pl. Zamkowym, stanął kontener, do którego przez 3 dni ustawiała się kolejka kilkuset osób, które stały w deszczu i w chłodzie, bo bardzo chciały się zaszczepić, bardzo chciały uratować życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych, uchronić przed potencjalnym zachorowaniem.

Ale szczepionki nie przyjechały do tej zamkniętej, ciepłej hali, w której ludzie mogą usiąść na krzesłach i bez kapiącego na głowę deszczu, w cieple poczekać na swoją kolej do szczepienia, tylko szczepionki przyjechały do oddalonego od tego miejsca o 2 km kontenera, do którego w kolejce ludzie musieli stać na dworze, w chłodzie, w deszczu, po kilka godzin dziennie. Pytam więc, dlaczego tak się dzieje. Nasuwa się tylko jedna odpowiedź: bo dla tego rządu ważniejsza jest propaganda niż szacunek dla zwykłego człowieka. Dziękuję. Doskonale pan, panie pośle, wie, że nie musieli. Były to dodatkowe możliwości zaszczepienia się. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ale również chciałbym się zwrócić do prezesa Rady Ministrów. Ptasia grypa, jak już powiedział pan poseł Ziejewski, zbiera bardzo duże żniwo w stadach, które są utrzymywane przez producentów drobiu.

W samym tylko powiecie kaliskim w Wielkopolsce - 55 ognisk. Oczywiście hodowcy, którzy mieli zakażone stada, musieli je utrzymywać, karmić, ponosić jeszcze dodatkowe koszty. Jest to dramatyczna sytuacja.

Jest największym eksporterem, wyprzedziliśmy tutaj Francję. Ta sytuacja może doprowadzić do załamania tej produkcji. Konieczne jest przede wszystkim pilne zwiększenie środków na wykupy, właściwie na zapłacenie odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z utylizacją stad. To są ogromne pieniądze w wypadku wielu producentów. Ponadto próba zwiększenia czy apele o zwiększenie tej kwoty adresowane do ministra rolnictwa spotykają się z odpowiedzią dla posłów, że w tej sprawie nie ma pozytywnej odpowiedzi ministra finansów. I to jest zadanie dla prezesa Rady Ministrów, do którego się zwracam, aby ta sprawa stała się ważnym punktem posiedzenia i decyzji rządu, żeby te pieniądze na odszkodowania były. Wielokrotnie z tej trybuny mówiłem o tym, że ta inspekcja ma ogromne potrzeby kadrowe, finansowe, ale również nieraz w sytuacjach, gdy trzeba pracować na okrągły zegar, umownie mówiąc, czyli 24 godziny, kiedy jest proces utylizacji tych stad, nie ma możliwości, aby pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej zapłacić za ponadnormatywne czasy pracy, ponieważ są oni pracownikami służby cywilnej.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Czesław Banot od wczesnego dzieciństwa związany był ze sportem. Już w wieku 10 lat rozpoczął treningi w klubie Piast Cieszyn, dla którego wywalczył awans do III ligi.

Wypadek na boisku w 1989 r. przerwał jednak jego działalność sportowo-szkoleniową. Po wypadku i częściowym paraliżu kończyn dolnych w ramach rehabilitacji zaczęła się jego przygoda z pływaniem. Od 1996 r. jako pływak niepełnosprawny znów aktywnie brał udział w zawodach sportowych, tym razem jako zawodnik niepełnosprawny Startu Bielsko-Biała, dla którego zdobył kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Czesław Banot to ikona samorządu Śląska Cieszyńskiego. Od 2006 r. do dnia śmierci nieprzerwanie pełnił funkcję radnego miasta Cieszyna, gdzie w sposób szczególny zabiegał o sprawy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, najmłodszych mieszkańców miasta, sportowców i rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego. Na zawsze, Czesławie, zostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ziemie wschodnich województw II Rzeczypospolitej zostały szczególnie doświadczone w okresie II wojny światowej. Na ludności tych terenów wywarły piętno dwa największe totalitaryzmy XX w. - narodowosocjalistyczna III Rzesza, Niemcy, i komunistyczny Związek Radziecki. Działania niemieckich i sowieckich okupantów stworzyły warunki do budzenia się nienawiści na tle narodowościowym ze strony Litwinów wobec Polaków oraz Żydów. Największej zbrodni na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej dokonano w miejscowości Ponary k. Wilna. Przygotowane w lesie przez sowietów doły dla planowanej bazy paliw Oddalenie Ponar od Wilna, a zarazem bliskość linii kolejowej i szosy pozwalały na sprawny transport osób przeznaczonych do zagłady. Niemcy wraz z kolaborującymi z nimi Litwinami ze specjalnego oddziału rekrutującego się ze Związku Strzelców Litewskich, zwanymi szaulisami, zamordowali w Ponarach ponad 100 tys. osób. W lesie ponarskim zginęła praktycznie cała diaspora żydowska Wileńszczyzny, ok. 70 tys. osób. Dokładna liczba zamordowanych Polaków ze względu na zatarcie przez okupantów śladów zbrodni nie jest niestety znana. Szacuje się, że w Ponarach zamordowano od kilku do kilkunastu, a nawet do 20 tys. Polaków. Obok Żydów i Polaków zginęli tam również jeńcy sowieccy, Białorusini, Romowie oraz Litwini. W Ponarach zgładzono polską elitę Wileńszczyzny, warstwę przywódczą narodu, żołnierzy ZWZ-AK, duchowieństwo, profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, nauczycieli, harcerzy, młodzież z konspiracyjnej organizacji Związek Wolnych Polaków. Przez zamordowaniem Polacy przychodzili ciężkie tortury w budynku gestapo przy ul. Ofiarnej oraz w więzieniu na Łukiszkach. Za kilka dni będzie kolejna rocznica tej zbrodni. W związku z tym apeluję o godne uczczenie ofiar tego mordu. Składam jednocześnie podziękowanie Kresowianom i ich potomkom, szczególnie członkom Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy i godnego upamiętnienia ofiar zbrodni w Ponarach. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Przede mną występowali posłowie, wygłaszając oświadczenia.

Szczególnie w tym dniu pamiętamy o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Druhny i druhowie, dziękuję wam za waszą służbę. Ślę moje najlepsze życzenia tylu powrotów, ile wyjazdów na akcje. Jako wiceprzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków życzę wam zdrowia, wielu przyjaciół. Dziękuję również waszym rodzinom. Oprócz tych życzeń życzę wam, aby rządzący chcieli wreszcie zająć się obywatelskim projektem ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników, dla rzeszy 500 tys. strażaków ochotników. Ten projekt leży już drugą kadencję. To dodatek w wysokości 300 zł za 20 lat służby, udział w akcjach. To nie ten projekt ustawy, o którym mówi rząd. Skromne pieniądze i podwyższenie lat służby. Bez was 40 tys. strażaków Państwowej Straży Pożarnej nie byłoby w stanie uczestniczyć w bardzo wielu akcjach.

Skierowaliście go do komisji. Przyjęcie tego projektu będzie najlepszym prezentem z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka dla tych, którzy poświęcają swoje życie, biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, którzy pod sztandarem: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek nie zważają na to, jakie zagrożenia na nich czyhają. To będzie odpowiedź i to będzie najlepszy prezent. Drugą kadencję leży ten projekt ustawy. To, co pochodzi od środowisk strażaków ochotników, powinno być uszanowane, jeśli mamy dla nich szacunek. Jeszcze raz: niech św. Florian ma was w opiece. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Niech św. Florian otacza was opieką, chroni od niebezpieczeństw.

Dziękuję za umożliwienie wygłoszenia dzisiaj oświadczenia. Pani Marszałek! Szanowna Izbo! Zostałam trochę sprowokowana, żeby tutaj wystąpić i wygłosić to oświadczenie, wypowiedziami niektórych posłów opozycji, którzy sugerują bardzo często w swoich wypowiedziach, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób uznaniowy kieruje środki finansowe do poszczególnych samorządów. Otóż, szanowni państwo, najlepszym przykładem tego, jak od lat środki finansowe były uznaniowo kierowane do poszczególnych samorządów, jest samo Mazowsze. Otóż w roku 2004, kiedy zdecydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej, wielu mieszkańców Mazowsza miało ogromne nadzieje na to, że te ogromne różnice, jakie są na Mazowszu, zostaną zniwelowane. Proszę państwa, przez wiele lat, przez te wszystkie lata, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, polityka, jaka jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, niestety doprowadziła do tego, że w roku 2018 doszło do wydzielenia NUTS 1 i NUTS 2, czyli tak jakby dwóch obszarów, właśnie z powodu ogromnego pogłębienia się różnic rozwojowych. Środki, które przez te wszystkie lata miały służyć zrównoważonemu rozwojowi. Wręcz przeciwnie, tak były one wydatkowane, że pogłębiły dysproporcje w rozwoju. Dlatego, proszę państwa, uważam - za to bardzo serdecznie dziękuję - że od 5 lat polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości służy właśnie nadrobieniu tych ogromnych zapóźnień.

Bardzo często powtarzam takie zdanie: dla niektórych włodarzy, patrząc na dane makroekonomiczne,

Dzisiaj dziękuję rządowi za to, że nadrabia to, czego niestety nie robią czy nie zrobili samorządowcy urzędu marszałkowskiego z Warszawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 29. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny kolejnego posiedzenia Sejmu, zwołanego na dni 19, 20 i 21 maja 2021 r., został paniom i panom posłom doręczony.